W dniu dzisiejszym, szanowni państwo, odbędzie się również posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To posiedzenie będzie miało miejsce od godz. 15.30. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Wysoka Izbo!

Pan dużo podróżuje w ostatnim czasie, ale chyba pan nie zauważył, że dzisiaj mamy 526 ofiar. To są kolejne istnienia ludzkie, które macie na sumieniu tylko dlatego, że nie prezentujecie żadnej spójnej strategii. Potraficie dużo mówić, ale nie jesteście w stanie wdrożyć rekomendacji własnej Rady Medycznej. Czas się skończył. Panie premierze, to już nie jest czas na to, byście prezentowali kolejne PR-owskie zagrywki. Czas wreszcie posłuchać ekspertów. Jest pan odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo wewnętrzne, ale również za zdrowie i życie Polaków. To nie był wniosek formalny. Pan poseł Wojciech Maksymowicz. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otóż gdybyśmy wprowadzili teraz obostrzenia, to wychodziłby pan Budka tutaj, na tę mównicę i mówił, że one są niepotrzebne. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Maksymowicz, Polska 2050. Proszę z wnioskiem formalnym, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przy okazji chciałem spytać panią marszałek, co się stało z poselskim projektem podobnej ustawy. Straty ludzkie są iście wojenne.

Ponieważ został złożony wniosek o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Z wnioskiem formalnym pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy składam wniosek formalny o odroczenie obrad do czasu przedstawienia przez premiera Morawieckiego i przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę informacji o wynikach śledztwa w sprawie domniemanego przestępstwa popełnionego przez wiceministra rządu ministra Łukasza Mejzę.

Chodzi o żerowanie na osobach chorych, umierających, niepełnosprawnych.

Po drugie, pan poseł Mejza złożył oświadczenie majątkowe. Ponieważ padł wniosek o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Proszę. Wysoka Izbo! 25 listopada pan minister Adam Niedzielski powiedział: Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu epidemii. 29 listopada, 4 dni później, pan minister wyszedł na konferencję prasową i poinformował o nowych obostrzeniach. Chcielibyśmy wiedzieć, kogo postawić przed sądem, czy tego ministra, który mówi w czwartek, że obostrzenia nie działają. czy tego, który w poniedziałek wprowadza te obostrzenia. To jest absurd, szanowni państwo.

Trzeba to jasno powiedzieć. Panie pośle, dziękuję bardzo.

Proszę panów o założenie maseczek.

Proszę o założenie maseczek. Obu panom posłom zwracam uwagę, że zakłócają panowie obrady Sejmu.

Obu panów na podstawie art. 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję do porządku i stwierdzam, że uniemożliwiają panowie prowadzenie obrad. Proszę o założenie maseczek. Pan poseł Grzegorz Braun oraz pan poseł Jakub Kulesza nadal uniemożliwiają prowadzenie obrad. Na podstawie art. 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu panów z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1793) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie!

Marszałek Sejmu skierowała uchwałę Senatu do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 26 listopada tego roku w celu rozpatrzenia. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu ośmiu poprawek na posiedzeniu 29 listopada wnosi, aby Wysoki Sejm wszystkie osiem poprawek odrzucił. W tym punkcie porządku dziennego głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Głosowało 430 posłów.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Senat zgłosił do art. 3 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw. Ogłaszam 2 minuty przerwy. Na tym zakończyliśmy głosowania.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wyrobach winiarskich (druki nr 1314 i 1776) Bardzo proszę panią poseł Teresę Pamułę o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, pani poseł.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów Publicznych wobec rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich, druki nr 1314 i 1776. Sejm na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu skierował do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komisji Finansów Publicznych projekt rządowy. Na wspólnym posiedzeniu wspomnianych komisji, które odbyło się w dniu 21 lipca br., została powołana podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich.

Na ostatnim posiedzeniu podkomisji w dniu 15 listopada 2021 r. zostało przyjętych 15 poprawek poselskich, które są wynikiem komentarzy Unii Europejskiej zgłoszonych w ramach notyfikacji oraz dyskusji w podkomisji, które z kolei wynikały z szerokiej konsultacji ze stroną społeczną, tj. organizacjami społecznymi zrzeszającymi producentów wina oraz fermentowanych napojów winiarskich, jak i uczelniami wyższymi. Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy dostosowania polskiego prawa do nowych przepisów odnoszących się do wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii Europejskiej, ujednolicenia wymagań dotyczących wpisu do rejestru działalności regulowanej, tj. rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich, i przyjmuje większość przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę po raz drugi.

Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich jest nową, kompleksową ustawą, która przyjmuje większość przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie, rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej oraz ujednolica i upraszcza wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej, rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Zaproponowane zmiany zmniejszają obciążenia administracji oraz usprawniają obieg dokumentów, co pozytywnie wpłynie na sytuację producentów, którzy chcą rozpocząć produkcję wyrobów winiarskich w Polsce. Projektowane przepisy przewidują wydanie czterech rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Na podstawie obecnych przepisów wydano osiem takich rozporządzeń. Najważniejsze rozwiązania to: zwiększenie konkurencyjności drobnych producentów wyrabiających cydr: cydr jakościowy, cydr lodowy, perry: perry jakościowe, perry lodowe, wina owocowe jakościowe oraz miód pitny jakościowy z surowców wyrabianych głównie we własnym gospodarstwie przy zwiększeniu maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów z 10 tys. l na rok do 100 tys. l na rok; umożliwienie produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni pszczelich; umożliwienie zakupu, do 50% pod względem wagowym, surowców do wyrobu takich napojów w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, lub w powiatach sąsiadujących z tym województwem; umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym; zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym, umożliwienie sprzedaży takich napojów w miejscu produkcji; zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów - to jest poprawka poselska. Ujednolicono przepisy dotyczące wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich. Podniesiono również wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich.

Uproszczono zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich. Dyrektor generalny KOWR będzie umieszczał wzór wniosku na stronach internetowych urzędu. Utworzono system elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami kontrolnymi w ramach sektora wina. Uproszczono system certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego.

Wprowadzono zezwolenia wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej w celu zniesienia barier administracyjnych, w tym tych związanych z obowiązkiem przekazywania jedynie najistotniejszych danych statystycznych dotyczących rynku wina. Warto również dodać, że rządowy projekt ustawy o wyrobach winiarskich był szeroko konsultowany ze stroną społeczną, tj. organizacjami społecznymi zrzeszającymi producentów wina oraz fermentowanych napojów winiarskich, jak również uczelniami wyższymi. Wysoka Izbo! Informuję, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierał rządowy projekt ustawy o wyrobach winiarskich w dalszych pracach legislacyjnych, Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę panią poseł Krystynę Sibińską, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jest to zupełnie nowa ustawa.

Ta ustawa jest oczekiwana przez środowisko winiarzy w Rzeczypospolitej, które jest dosyć liczne, bo przypomnę tylko, że zgodnie z danymi gromadzonymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarejestrowanych jest 329 producentów wina. Dotyczy to rzeczywiście wielu działalności, o czym rozmawialiśmy i nad czym procedowaliśmy w trakcie prac zarówno podkomisji, jak i komisji. Rzeczywiście proponowana ustawa wprowadza bardzo dużo zmian. Chodzi o zakres wyrobu fermentowanych napojów winiarskich. Upraszcza, ujednolica zapisy.

Ogranicza dużo takich procedur administracyjnych, aczkolwiek nie wszystkie, o tym będę mówiła w dalszej części wystąpienia.

Podkomisja zbierała się kilkakrotnie.

W tym momencie bardzo dziękuję lubuskim winiarzom, z którymi miałam przyjemność się spotkać, wymienić uwagami. Niektóre z nich zostały uwzględnione w czasie prac podkomisji, za co też dziękuję. Tak że rzeczywiście prace nad tym projektem rządowym były bardzo, bardzo poprawne, jeśli chodzi o proces legislacyjny. Myślę, że głosowanie pokaże, że w taki sposób procedowana ustawa może przejść niemalże jednogłośnie, tak jak się zdarzyło na połączonych posiedzeniach komisji rolnictwa i Komisji Finansów Publicznych. Mianowicie winiarze zgłaszali np. taką uwagę, że niektóre terminy są niepowiązane z kalendarzem winiarskim i wypadają wtedy, kiedy oni są najbardziej zapracowani.

Udało się wprowadzić dwie poprawki, które umożliwiają drobnym producentom wina i rolnikom, którzy też produkują wyroby winiarskie, sprzedaż bezpośrednio do restauracji, do barów, do lokalnych sklepów. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że to jest też promocja (Dzwonek) lokalnych wyrobów. Jedna rzecz, o której należy wspomnieć, mianowicie: sprawa związana z akcyzą.

Natomiast jest to związane z tym, że w Europie nie ma takich przepisów. Zarówno w pracach podkomisji, jak i komisji apelowaliśmy do komisarza do spraw rolnictwa. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem tych przepisów.

Zapraszam, panie pośle. Dzień dobry. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie projektu ustawy o wyrobach winiarskich zawartego w druku nr 1314. Rzeczywiście jest to ustawa, która przez całą branżę była długo oczekiwana, bo widać wyraźnie, że rozwija się przemysł winiarski w Polsce. Oczywiście pewnie daleko nam jeszcze do takich krajów jak Hiszpania, Portugalia, Francja czy Włochy, które rzeczywiście są potęgą, jeżeli chodzi o produkcję win. Natomiast ta ustawa wprowadza rozwiązania podobne do tych, które funkcjonują w krajach Unii Europejskiej, i daje możliwość rozwoju całej branży.

Ustawa również porządkuje wiele przepisów, które do tej pory były bardzo niejasne i powodowały trudności interpretacyjne.

Co to powoduje? Otóż przede wszystkim poprawia się sytuacja właśnie drobnych producentów win, cydrów, win owocowych, miodów pitnych. Na podstawie tej ustawy, jeżeli ona zostanie przyjęta, zdecydowanie łatwiej będzie można taką działalność rozpoczynać.

Oczywiście w Polsce na ten moment mamy 230 producentów win i zaledwie kilku, którzy ten próg przekraczają, w związku z czym niewątpliwie jest to szansa na rozwój dodatkowych podmiotów, tworzenie nowych miejsc pracy i niewątpliwie doprowadzi to do rozwoju lokalnych producentów. Ustawa, i to są bardzo dobre zapisy, reguluje kwestie procedur związanych z produkcją tych napojów, z produkcją win. Wreszcie będzie wprowadzana ewidencja winnic.

To jest też bardzo istotna sprawa i istotna zmiana.

To też jest bardzo dobre rozwiązanie, które niewątpliwie pobudzi również funkcjonowanie tego rynku w Polsce. Oczywiście w tym wszystkim bardzo ważną rzeczą są kwestie związane z akcyzą, z rozliczeniem podatkowym, jeżeli chodzi o produkcję win, cydrów, win owocowych.

Reasumując, klub Lewicy (Dzwonek), będzie głosował za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pan poseł Jacek Tomczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego PSL - Koalicja Polska w związku ze sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wyrobach winiarskich, druk nr 1314. Niewątpliwie przyszłość i rozwój polskiego rynku winiarskiego winny być przedmiotem troski władz publicznych, w tym troski polskiego ustawodawcy. Rozwój sektora polskiego rolnictwa i przetwórstwa stanowi istotny element wzmacniania całej gospodarki.

Polscy producenci wina, cydru, perry czy miodów pitnych bez kompleksów stają również do jakościowej konkurencji z producentami z innych krajów.

Ustawa wprowadza także zasady znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie ich nazw przewidzianych prawem zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Istotnych zmian jest znacznie więcej, mamy szereg ułatwień administracyjnych.

Już dzisiaj wiadomo, że w tym projekcie nie ma zapisu zezwalającego na to, żeby restaurator, który chce sprzedać obiad, mógł dołożyć do tego obiadu butelkę producenta polskiego wina. A więc niektóre regulacje są zdecydowanie za wąskie.

Mogą je oferować przez Internet firmy zagraniczne poza naszymi granicami. Nie mogą ich oferować niestety polscy producenci win. Ta ustawa tylko ułatwia sprzedaż producentom.

Większość krajów unijnych w trakcie pandemii zniosła wszelkie zakazy, limity. To jest niezrozumiałe (Dzwonek), bo podwyższamy opłatę i utrudniamy sprzedaż polskich alkoholi przez Internet.

Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękujemy za poprawkę. Zapraszam.

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce.

Większość polskich konsumentów bardzo mocno to odczuje. Przypomnę, że mówimy o samych podatkach, a nie możemy też zapomnieć o rosnącej inflacji, w przypadku której niby jest jakaś propozycja, ale powoli już przestajemy w to wierzyć, bo ta hipokryzja jest ogromna. Szanowni państwo, przypomnę też, że rząd nie przewiduje przeznaczania tych środków de facto na działania profilaktyczne, więc jest to tylko i wyłącznie ordynarne strzyżenie portfeli Polaków. Popieramy tę ustawę.

Jest to krok w dobrą stronę, ale to nie ukryje całej masy innych utrudnień, które państwo już Polakom zgotowali, takich jak choćby segregacja sanitarna. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Koło Parlamentarne Polska 2050 oczywiście będzie głosowało za tym projektem, za tą ustawą. To jest dobra ustawa. Ta ustawa sama w sobie jest oczywiście pochodną ustawodawstwa Unii Europejskiej, ale cieszy w wielu różnych aspektach, z których większość została już poruszona. Odniosę się tylko do dwóch, może trzech. Bardzo cieszy zwiększenie konkurencyjności drobnych producentów cydrów, pitnych miodów czy win owocowych wytwarzanych z surowców we własnych gospodarstwach. Istotne dla nas - nie tylko dla nas, głównie dla rynku - jest zróżnicowanie segmentów cydru i perry, gdzie oprócz standardowych produktów pojawiają się produkty jakościowe. To istotna dla branży winiarskiej zmiana, choćby dlatego, że za granicą popularność tego rodzaju wyrobów z roku na rok rośnie.

To jest krok w dobrą stronę. W ten sposób polski Sejm zaczyna się jawić jako zagłębie analogowej korespondencji, jedno z ostatnich w naszym kraju. To bardzo niedobrze. Na poprzednim etapie akcentowaliśmy potrzebę harmonizacji projektowanej ustawy z przepisami, które regulują pobór akcyzy. Temu wyzwaniu też niestety nie sprostano. Branża sygnalizuje potrzebę zaangażowania Ministerstwa Finansów w rozwiązanie tego problemu. Liczymy na to, że do takiego zaangażowania dojdzie. To przedłożenie wprawdzie nie otwiera drogi lokalnym producentom aż tak szeroko, jak np. ustawodawstwo kanadyjskie - znany jest kazus belgijskiego imigranta Pascala Miche, który najpierw udowodnił, że pomidory są owocami, a potem uzyskał oficjalne pozwolenie na produkcję wina z pomidorów - ale za to odnosi się wprost do tradycyjnego polskiego trunku, czyli miodów pitnych jakościowych. Jest to jeden z wielu elementów, dzięki którym koło Polska 2050 zagłosuje za tą ustawą. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, zgłosiło się 10 osób do zadania pytań. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Jest pan poseł Adamczyk? Pan poseł Jan Szopiński.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmierza się do tego, aby przedsiębiorca, u którego stwierdzono naruszenia warunków określonych w art. 8 ust. 1 lub 2, mógł usunąć te naruszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W związku z tym chciałem zapytać pana ministra o to, w jaki sposób te terminy będą określone. Może się okazać, że przy tak bardzo sztywnym i niezbyt proprzedsiębiorczym podejściu niektórych urzędów taki przedsiębiorca nie zdąży usunąć takich wad, co byłoby ze szkodą zarówno dla rynku, jak i dla samego przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Przedstawiciele Rządu! Wysoki Sejmie! Celem tej ustawy, jak już była mowa, jest przede wszystkim potrzeba dostosowania polskiego systemu prawnego do wszystkich aktualnie obowiązujących aktów unijnych.

Chciałbym zapytać. Jednym z celów ustawy, o których się mówi, jest nowy podział kompetencji organów kontrolnych. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku!

Mówiono także. Komisje, które zajmowały się tym problemem, to komisja rolnictwa i Komisja Finansów Publicznych. Ja natomiast oczekiwałabym, że ta ustawa jednak będzie skonsultowana z komisją społeczną i z organizacjami, które zajmują się przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Pan poseł Jacek Tomczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Polskie winiarstwo cały czas się rozwija, wymaga też wsparcia.

Natomiast żeby tak się stało, musimy otworzyć sprzedaż alkoholu przez Internet, tak żeby udrożnić kanały sprzedaży, umożliwić polskim producentom sprzedaż nie tylko tego, co wyprodukują w swojej siedzibie, w swojej winnicy, bo ten projekt dotyczy tylko tego elementu, ale także umożliwić restauratorom możliwość oferowania swoich dań z polskimi winami czy polskimi piwami, czy innymi jakościowymi trunkami. To otwarcie jest niezbędne.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Małgorzata Pępek, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Przytaczane spostrzeżenia dotyczące ustawy, jak również opinie przedstawicieli wytwórców bezpośrednio obecnych na sali pokazały, z jakimi problemami spotykają się producenci wyrobów winiarskich w praktyce. Często z pozoru błahe kwestie mają ogromne znaczenie i wpływ na zachowanie procesu przetwórstwa, jak również przysparzają problemów związanych z zachowaniem chociażby terminów urzędowych. Jest to niezwykle ważne, żeby wspierać polskich producentów. Chciałabym zapytać: Jakie dodatkowe działania podejmie rząd, aby promować i wspierać polskich producentów wyrobów winiarskich? Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam dwa konkretne pytania dotyczące procedowanej materii ustawowej.

Musimy pamiętać, że winiarstwo związane jest także z działalnością gospodarstw agroturystycznych czy też polskich restauratorów. Czy planujecie państwo pomoc, która byłaby adresowana do polskich winiarzy, w zakresie możliwości pozyskania areału ziemi, chociażby tej, która jest w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy jakieś preferencyjne ceny, czy sposób przekazywania polskim winiarzom gruntów? Drugi wątek, o którym chcę powiedzieć, to właśnie kwestia e-commerce, czyli dostępności polskiego wina produkowanego w granicach administracyjnych państwa polskiego dla polskich restauratorów, tak aby mogli oni zaopatrywać się, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemicznym, właśnie w sposób elektroniczny. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Według prognozy będzie to dotyczyć wielu podmiotów. Czy będzie to możliwe? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Beata Strzałka, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiany w ustawie były długo oczekiwane przez producentów win, nie tylko win jakościowych, ale także cydrów i perry, o czym świadczy właśnie szeroki udział w pracach komisji i podkomisji przedstawicieli branży winiarskiej. Zostały uporządkowane definicje i kategorie tych produktów, ale ustawa zawiera także zmiany dotyczące ilości win produkowanych przez właścicieli winnic, których bardzo dużo powstaje w Polsce i które wytwarzają dobre, jakościowe produkty.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke, koło Konfederacja.

Ja z miłości do pana posła. Dziękuję. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Konfederacja z zadowoleniem oczywiście wita tę ustawę, która poszerza swobody ludzi.

Były takie czasy, kiedy wymyślono samochody, i wtedy przed samochodem musiał biec chłopiec z czerwoną chorągiewką, ostrzegając ludzi. Po jakimś czasie te ograniczenia zlikwidowano. Dlaczego np. jedni mogą sprzedawać swoje wina bezpośrednio gdzieś w restauracji, a drudzy muszą poprzez hurtownie?

Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem zadać dwa pytania.

Bo czasami takie wina są w naszym kraju produkowane.

Pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przewrotnie zapytać: Czy podatek cukrowy jest naliczany również w przypadku napojów alkoholowych? Pragnę przypomnieć, że został on wprowadzony u nas pod pretekstem ochrony zdrowia Polaków. Czy litr wina dosładzanego identyczną ilością substancji słodzących podlega tym samym obciążeniom co litr innych napojów? Jeżeli tak się nie dzieje, to prosiłbym o wyjaśnienie, jakie zbawienne odziaływanie na ludzki organizm według twórców ustawy ma alkohol, jeśli neutralizuje tak szkodliwy cukier, ewentualnie jakie inne przesłanki wpłynęły na takie rozwiązania, chyba że przy wprowadzaniu podatku cukrowego nie chodziło o zdrowie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Nie ma pana posła. W takim razie przechodzimy do odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Norbert Kaczmarczyk wszystko to państwu wyjaśni. Zapraszam, panie ministrze.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy o wyrobach winiarskich jest niezwykły, jeżeli chodzi o prowadzenie go w parlamencie.

To dzięki temu wielkiemu konsensusowi i tej wielkiej, wspaniałej pracy całego parlamentu udało się doprowadzić projekt do takiego stanu.

Jedną z nich jest kwestia związana ze sprzedażą przez Internet. Muszę państwu powiedzieć, że jest to kompetencja Ministerstwa Zdrowia i jeżelibyśmy chcieli zmieniać w tym kontekście tę ustawę, to rzeczywiście jest to kompetencja resortu zdrowia. Oczywiście prace nad tym trwają.

Wielu z państwa parlamentarzystów pytało o tę kwestię, o dostępność przez Internet. To rzeczywiście byłoby rewolucyjne, jeżeli chodzi o nasz rynek. Natomiast te rozmowy pozostają otwarte. Natomiast dziękuję klubowi Koalicji Polskiej również za aprobowanie innych przepisów tej ustawy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z pytaniami państwa posłów, to chociażby pan poseł Tadeusz Tomaszewski pytał o organy kontrolne.

Natomiast pani poseł Joanna Fabisiak pytała o polski produkt, profilaktykę, czyli kwestię związaną z wychowaniem w trzeźwości. Właśnie tutaj jest sprzeczność, bo z jednej strony niektórzy z państwa chcieliby sprzedaży przez Internet, a z drugiej strony inni parlamentarzyści pytają o profilaktykę. Profilaktyka na dzisiaj funkcjonuje na starych zasadach, więc jeżeli mielibyśmy wychodzić naprzeciw konsumentom i sprzedawać przez Internet te wyroby alkoholowe, to musimy zastanowić się nad mocną profilaktyką. Wielu z państwa parlamentarzystów na etapie prac nad tą ustawą pytało również o reklamę, o to, dlaczego nie możemy reklamować alkoholu tego typu. Tutaj również kłania nam się ustawa o wychowaniu w trzeźwości i kompetencje Ministerstwa Zdrowia. Pan poseł Jacek Tomczak również pytał o sprzedaż alkoholu przez Internet. Mam nadzieję, że szczegółowo na temat tych planów będziemy mogli pani poseł odpowiedzieć na piśmie. Ta ustawa na pewno jest bardzo ważnym krokiem i konsensusem, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, jeżeli chodzi o zmniejszanie obciążeń administracyjnych, jeżeli chodzi o sprzedaż wyrobów winiarskich. Pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek pytała o sprzedaż, o wielkość sprzedaży w miejscu wytworzenia.

Ten projekt konsumuje to i zadowala osoby, które rzeczywiście będą się tą branżą zajmowały.

Oczywiście taka jest nasza rola. Również komisja do spraw deregulacji powstała po to, by te przepisy upraszczać. Natomiast ten przepis, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, jest bardzo ważny w porozumieniu z tym ostatnim projektem. Również jest on przyjęty w wielkim konsensusie, jeżeli chodzi o ustawę o sprzedaży w piątki i soboty przez rolników na lokalnych targowiskach, umożliwieniu im tego przez samorządowców. To bardzo ważny projekt, który w pewien sposób z tym koreluje.

To jest bardzo ciekawy temat. Na pewno chociażby Małopolska Hodowla Roślin czy inne instytuty chętnie podejmą ten temat.

Natomiast niektóre pomysły powinny pozostać podtrzymane, a nie poprzez tę, niestety, transformację wykonaną niekoniecznie w sposób adekwatny do warunków panujących w Polsce. Powinniśmy pewne pomysły przejąć, chociażby taki jak te instytuty, które budowały określone odmiany roślin dla określonych terenów. Pamiętam chociażby z moich terenów takie instytuty, jeżeli chodzi o budowę genetyki, jeżeli chodzi o tytoń i uwarunkowanie glebowe dla tych roślin, więc to jest niesamowicie istotne. Popieram ten argument, aby rozpocząć prace albo kontynuować to w miejscach, gdzie rzeczywiście te prace zostały rozpoczęte. Jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedziałem, to oczywiście odpowiemy na piśmie. Serdecznie dziękuję za tak dobre, mądre i spokojne procedowanie nad tą ustawą. Mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli tak dobrze pracować w parlamencie. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Myślę, że to akurat do tej dyskusji bardzo pasuje, bo picia wina i alkoholu, jak wiemy, nie należy zalecać. Woda - zdrowa.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym bardzo serdecznie właśnie stąd podziękować przewodniczącemu nadzwyczajnej podkomisji do spraw wyrobów winiarskich, bo to dzięki jego determinacji i współpracy pomiędzy rządem, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministerstwem finansów oraz Ministerstwem Zdrowia.

Dziękuję serdecznie. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Wysoka Izbo! Zwracam się do pana ministra z prośbą po raz wtóry. Otóż chciałabym prosić o przedstawienie informacji co do profilaktyki. Czy nie uważa pan, że wobec zwiększenia zakresu produkcji, co jest rzeczą dobrą, bo jest otwarcie dla przedsiębiorców, powinna być choćby informacja, że młodzieży, szczególnie młodzieży niepełnoletniej, wina się nie sprzedaje?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (druki nr 1694 i 1772) Proszę pana posła Kazimierza Chomę o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!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 Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r. wnoszą, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Chciałbym nadmienić, że projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych w grudniu 2020 r.

W ramach opiniowania projekt został skierowany do 21 podmiotów, m.in. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz marszałków poszczególnych województw. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostały poddane analizie i w znacznej części uwzględnione.

Projekt ustawy z poprawkami został jednogłośnie uchwalony przez połączone komisje. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Zapraszam pana posła Kazimierza Chomę z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, czyli tego samego klubu co przed chwilą, o zabranie głosu. Proszę bardzo.

Wysoka Izbo! Mam wielki zaszczyt w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości zaopiniować projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, druk nr 1694. Projekt ustawy wychodzi naprzeciw potrzebom usprawnienia oraz przyspieszenia procedury prowadzenia postępowań scaleniowych w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

Z analizy danych w tym zakresie dotyczących niektórych krajów Unii Europejskiej wynika, że wielkość ta wynosi w skali roku nawet do 3% powierzchni gruntów rolnych danego kraju, co w warunkach polskich oznaczałoby powierzchnię ok. 450 tys. ha rocznie.

Po pierwsze, reguluje się procedury postępowania w przypadku wprowadzenia na części albo na całym terytorium RP stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to realizowane dzięki możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji wszelkich zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. W ustawie rezygnuje się z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego, a także z podejmowania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia.

Po drugie, wprowadza się terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, co pozwoli na wykonanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych. Po trzecie, wprowadza się definicję gospodarstwa rolnego zawierającą szczególną normę obszarową, co upraszcza weryfikację wniosków o wykonanie scalenia gruntów. Po czwarte, doprecyzowuje się czynności związane z określeniem przebiegu granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów. Po piąte, włącza się przedstawiciela gminy oraz sołtysa do komisji doradczej. Po szóste, wskazuje się starostę jako organ właściwy do wnioskowania do sądu wieczystoksięgowego.

Po dziewiąte, upraszcza się sposób zamknięcia przez sąd księgi wieczystej w drodze czynności technicznej podejmowanej na skutek zawiadomienia właściwego starosty bez wydawania przez sąd postanowienia w tym zakresie. Jak widać z przedstawionej analizy, rządowy projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, druk nr 1694, jest bardzo potrzebny i klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za jego przyjęciem.

Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koalicja Obywatelska po przeanalizowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych uznaje, że proces wymiany i scalenia gruntów jest konieczny i bardzo potrzebny. Wynika to z konieczności ustalenia m.in. stanu prawnego gruntów. Jednakże niektóre zapisy tej ustawy wymagają wyjaśnienia.

Gospodarstwa te powstaną w wyniku scalenia gruntów rolnych i leśnych. O ile zwiększy się powierzchnia gruntów w Polsce objętych płatnościami bezpośrednimi? Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że w warunkach polskich ok. 450 tys. ha gruntów rocznie miałoby podlegać scaleniu. To wynika z danych dotyczących niektórych państw Unii Europejskiej, gdzie ok. 3% powierzchni gruntów rolnych podlega scaleniu.

150 lat. Panie Ministrze! Czy rząd wobec tak ambitnego programu scaleń jest wystarczająco przygotowany pod względem organizacyjnym i finansowym, aby wykonać plan scaleń? W ocenie skutków regulacji napisano, że wdrożenie tego programu nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie ponosił koszty wdrożenia tej ustawy w życie. Naszym zdaniem koszty będą po stronie administracji rządowej, samorządowej, jednostek geodezji i sądów. W tym projekcie tych kosztów nie wykazano. W projekcie ustawy jest zapis nakładający na sądy administracyjne rozpatrzenie skargi w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów w terminie 2 miesięcy.

Panie ministrze, czy w sądach administracyjnych będą stosowne procedury, które spowodują przyspieszenie wydawania decyzji zgodnie z zaleceniem ustawodawcy?

Zadanie jest bardzo, bardzo trudne.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Romuald Ajchler, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Lewica popiera projekt ustawy. Uważamy, że zmiany zawarte w projekcie poprawią proces wymiany i scalania gruntów, a także usprawnią ten proces. Jest szansa na to, że go w znaczący sposób skrócą. Ta ustawa wychodzi naprzeciw tym problemom, które były dostrzegane w przypadku scalania i wymiany gruntów na podstawie starej ustawy. Ale jest jedno „ale”, Wysoka Izbo. Myślę tu o rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i ich członkach.

Dochodzi do takiej sytuacji, że jeżeli członek spółdzielni chce grunty wymienić ze spółdzielnią, natychmiast może wejść firma państwowa i te grunty przejąć. Uważamy, że rząd powinien nad tą sprawą się pochylić i doprowadzić do oczywistej rzeczy. Dzisiaj wielu członków spółdzielni odchodzi na emeryturę i chce pozostawić te grunty w spółdzielni, w jej użytkowaniu. Nie ma takiej możliwości, bo nawet gdyby chcieli sprzedać te grunty spółdzielni, te grunty są przejmowane przez ARiMR. Wysoka Izbo! Projekt ustawy nie wzbudził kontrowersji. Nie było żadnych merytorycznych poprawek, jeśli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem, z wymianą gruntów. Posłowie i komisje doszli do wniosku, że ta ustawa idzie w dobrym kierunku i pomoże rolnikom w procesie wymiany tych gruntów. Powtarzam jeszcze raz, że należałoby się przyjrzeć Prawo spółdzielcze w kontekście wymiany gruntów pomiędzy podmiotami pracującymi w spółdzielni, a także samym spółdzielniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, druki nr 1694 i 1772. Scalanie gruntów jest fundamentalnym zabiegiem w procesie urządzania przestrzeni wiejskiej przyczyniającym się do wyeliminowania barier rozwojowych danej wsi poprzez likwidację wadliwej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie scaleniowe niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, rozpoczynając od starosty, który po zrealizowaniu procedury będzie miał uporządkowaną bazę danych w przypadku ewidencji gruntów i budynków, przez wójta, który poza wydzieleniem rezerwy terenowej pod grunty miejscowej użyteczności publicznej skorzysta z przeprowadzonego zagospodarowania poscaleniowego w postaci zmodernizowanej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, a kończąc na rolnikach, którzy w rezultacie będą kompletnymi beneficjentami tego przedsięwzięcia i otrzymają jedyną w swoim rodzaju szansę na podwyższenie efektywności prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych.

Scalenie gruntów daje również możliwość realizacji zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na danym obszarze, także w zakresie małej retencji wodnej, oraz zadań wpływających na poprawę walorów estetycznych krajobrazu rolniczego.

Ta sytuacja pandemiczna spowodowała to, że nastąpiły opóźnienia, bo chociażby zwołanie zebrania wiejskiego, na którym ogłaszano informacje dotyczące postępu prac scaleniowych, było niemożliwe. W związku z tym i wojewódzkie biura geodezji, i samorządy zgłaszały uwagi, że trzeba w końcu podjąć decyzję, by wykorzystać możliwości internetowe, by zamieszczać informacje w Biuletynie Informacji Publicznej, bo te informacje mogą być ogólnodostępne, a problem pojawiał się, kiedy na spotkanie przychodziło 3–4 mieszkańców danej miejscowości czy uczestników scalenia, a do reszty trzeba było docierać.

Na to też czekali mieszkańcy terenów objętych scaleniami. Trzeba dokonać tych zmian, żeby przepisy wynikające z ewidencji gruntów i budynków i to, co jest zawarte w księgach wieczystych, były ze sobą spójne, żeby współgrały. Jeżeli tych zmian byśmy nie wprowadzili, te procesy będą się przedłużać. Wszystkie proponowane rozwiązania przyczynią się do usprawnienia procesu, jakim jest scalanie gruntów, i spowodują jego sprawną realizację, a tym samym umożliwią wojewódzkim biurom geodezji oraz starostom realizację większej liczby projektów, na które czekają rolnicy w całym kraju, bo to nie tylko scalanie gruntów, ale to też te całe procesy poscaleniowe, które regulują gospodarkę, ułatwiają wymianę gruntów, dają możliwość uregulowania bez aktu notarialnego sytuacji prawnej wielu gospodarstw. Jest to działanie ze wszech miar potrzebne i oby sprawniej, oby szybciej, oby więcej (Dzwonek) udało nam się zrobić. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku!

Już za 2 tygodnie pokażą to w Brukseli, gdy 13 grudnia wraz z rolnikami z całej Europy powiedzą zdecydowane „nie” dla Europejskiego Zielonego Ładu, a właściwie nieładu, który doprowadzi do zapaści polskiego i ogólnoeuropejskiego rolnictwa. Pseudoekologiczni zieloni fanatycy z Unii Europejskiej w imię neutralności klimatycznej doprowadzą do sytuacji, w której europejscy rolnicy przestaną się liczyć zarówno na rynku krajowym czy rynku wewnętrznym, jak i na rynkach światowych, w handlu międzynarodowym. Unia Europejska może doprowadzić do sytuacji, w której ceny żywności gwałtownie wzrosną, a nasze rynki po prostu zostaną zalane przez produktu z innych kontynentów. Likwidacja chowu klatkowego, ograniczenie wykorzystania areałów ziemi, które też jest zapowiadane. Drastycznie wpłynie to na wydajność właśnie tego polskiego, ale i europejskiego rolnictwa, tej produkcji, a wartość eksportu po prostu spadnie. Takie działania doprowadzą do tego, że do Europy trafi po prostu więcej importowanej żywności. Zastanawiam się, czy to jest właśnie celem eurokratów, czy zubożenie polskiego rolnika i skazanie Polaków na żywność z importu to jest cel eurokratów i tych tzw. ekologów z Unii Europejskiej. Dziś jako politycy powinniśmy solidarnie z rolnikami wyrzucić Europejski Zielony Ład tam, gdzie jest jego miejsce - na śmietnik. Miejmy nadzieję, że na tym samym śmietniku historii skończą też pomysłodawcy, autorzy tych szalonych pomysłów. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pani posłanka Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa nie budzi wątpliwości, ona jest korzystna, my ją oczywiście poprzemy.

A więc to jest nie tylko kwestia wiejska, ale też jak najbardziej kwestia miast. Koło Parlamentarne Polska 2050 składa dwie poprawki. W tym projekcie wprowadza się niezwykle krótki termin 2-letni, po upływie którego nie będzie możliwości uchylenia decyzji administracyjnej. Mając na względzie realne zapewnienie stronie postępowania prawa do sądu oraz uwzględniając stan epidemii, projektowany termin będzie oznaczał znaczące ograniczenie prawa strony do wzruszenia decyzji administracyjnej.

Druga poprawka mówi o tym, co nie zasługuje na naszą aprobatę, a mianowicie o proponowanym wprowadzeniu specjalnych terminów rozpatrzenia skargi w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów. W praktyce przedmiotowy termin będzie niemożliwy do spełnienia przez Sąd Administracyjny. Z uwagi na trwający stan epidemii już teraz rozpatrzenie sprawy przed Sądem Administracyjnym w terminie 2 miesięcy jest terminem nierealnym, tym samym nierozpatrzenie sprawy w tym terminie będzie automatycznie stwierdzeniem naruszenia prawa. Z tego względu proponujemy wprowadzenie tych dwóch poprawek, które w tej chwili panu marszałkowi przekazuję. Proszę państwa, przechodzimy do zadawania pytań. Dziewięć osób zgłosiło się do zadania pytań. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Pan poseł nie wrócił.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moi wyborcy pytają, czy dzięki temu rozwiązaniu zbyt aktywnego, protestującego przeciwko władzy rolnika władza ta za pośrednictwem starostów będzie miała prawo przenieść na drugi kraniec Polski. To przekazuję, bo takie otrzymałem pytanie. Proszę też o wytłumaczenie, w jaki sposób w majestacie prawa można przerwać postępowanie spadkowe i uniemożliwić spadkobiercy objęcie spadku lub narzucić mu wymianę tego spadku na inny, w sytuacji gdy wartość masy spadkowej nie została oszacowana przez stronę, gdy toczą się jeszcze spory pomiędzy spadkobiercami.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Wysoka Izbo!

Dlaczego cała procedura trwa tak długo? Czy oprócz proponowanych przez rząd rozwiązań nie można uprościć tej procedury jeszcze bardziej? Chciałabym też zapytać, jak wygląda sytuacja w województwie pomorskim związana właśnie ze scalaniem i wymianą gruntów. Jak duży jest to problem i kiedy działki chętnych właścicieli zostaną scalone?

To będzie naprawdę skomplikowana procedura.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mimo że niektórzy nie mogą tego przyjąć do wiadomości, to nasz świat stoi na progu klimatycznej katastrofy. Najbardziej odczuwają to rolnicy, którzy już teraz ponoszą straty i cierpią z powodu nagłych zmian pogodowych. Uważam, że zmiana art. 1 poprzez zaakcentowanie nowego celu scalania, którym jest zabezpieczenie gruntów przed ich degradacją klimatyczną, jest trafna. Rząd po prostu ucieka od problemu. Skoro podczas konsultacji pojawiają się uwagi i wątpliwości, to oznacza, że istnieje konieczność podjęcia dyskusji i dokonania pogłębionej analizy sygnalizowanych rozwiązań i ustawowe ich wdrożenie. Mądry rząd to taki, który jest mądrością innych, w tym przypadku specjalistów. Czy ministerstwo w toku prac nad tym projektem zamierza uwzględnić nowelizację art. 1 z uwagami zgłoszonymi przez środowiska naukowe - Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów i Stowarzyszenia Geodetów Polskich? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze!

Termin został określony na co najmniej 7 dni przed terminem podjęcia czynności, termin wykonania tej czynności. Chciałem zapytać, czy to nie jest jednak zbyt krótki czas, ponieważ bardzo często jest to związane z obowiązkami. Zwolnienie się i uczestnictwo w takiej procedurze jest związane z koniecznością odstąpienia od obowiązków zawodowych czy też innych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę. Wysoka Izbo! Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań scaleniowych jest rozwiązaniem potrzebnym. Trwająca pandemia dowiodła, że podobnie jak w przypadku np. Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do możliwości zdalnego procedowania przez organy spółek muszą istnieć normy pozwalające na przeprowadzenie scaleń niezależnie od trwającej pandemii. Słuszne uwagi budzi czas tej nowelizacji. Dlaczego dopiero po 2 latach od wybuchu epidemii wprowadzacie pod obrady ten projekt? Najbardziej fundamentalne dla państwa regulacje przepychaliście nocami z pogwałceniem wszelkich procedur, a na przepisy, które mogą realnie przysłużyć się obywatelom ze względu na trwającą pandemię, trzeba było czekać tyle czasu. Co jest powodem tak dużego opóźnienia? Pan poseł Tomasz Głogowski, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Przy okazji tego projektu ustawy dotyczącego scalania gruntów i funkcjonowania ksiąg wieczystych chciałem poruszyć problem czasu dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. On jest zróżnicowany w różnych miejscach, to zależy od sądu. A sensowny i sprawny termin dokonywania wpisu w księgach wieczystych jest ważną sprawą, jeśli chodzi o obrót gospodarczy, jest ważną sprawą dla gospodarki.

Opóźnienia w tej chwili wynikają przede wszystkim z braku odpowiedniej liczby referendarzy w odpowiednich wydziałach sądów. Czy ministerstwa mają tego świadomość i planują jakieś działania zmierzające do poprawy tej sytuacji? Dziękuję serdecznie. Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Chyba nie widzę pana posła. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub parlamentarny Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowni Przedstawiciele Rządu!

Tutaj dodaje się przedstawiciela gminy i przedstawiciela sołtysa lub przedstawiciela rady sołeckiej miejscowości, które objęte są programem, projektem scalania. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że ono może eliminować napięcia społeczne, zwłaszcza kiedy będzie to przedmiotem funkcjonowania tej komisji.

Chciałem zapytać przede wszystkim o to, jakie są przeznaczone na przyszły rok środki wynikające ze wsparcia scalania gruntów na przyszły rok i na kolejne lata. Po drugie, wiemy, że w przyszłym finansowaniu wspólnej polityki rolnej odbiera się urzędom marszałkowskim dysponowanie tym programem, który przez wiele lat się sprawdził. To urzędy marszałkowskie miały pełną infrastrukturę, a przede wszystkim osoby odpowiedzialne na poziomie regionalnym właśnie za scalanie gruntów. Trzecia rzecz: Jak wyglądają w podziale na województwa właśnie elementy scalania gruntów? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Krzysztof Ciecióra. Zapraszam serdecznie, panie ministrze.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wszystkim bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję.

Jest to ustawa, którą nowelizujemy.

Średnio, na podstawie danych statystycznych z poprzednich lat, koszt scaleń wynosił ok. 100 mln zł rocznie. Ponadto w nawiązaniu do tej nowelizacji i do przewidywań, że zainteresowanie scaleniami może wzrosnąć, mamy dodatkowo zagospodarowane, zabezpieczone 137 mln euro do 2027 r., czyli mamy skąd te pieniądze dodatkowo przesuwać w sytuacji, w której będzie taka potrzeba. Właśnie to jest kwota, która to wyczerpuje. Warto podkreślić, że to nie gminy prowadzą ten proces, tylko starostwa. Jeżeli chodzi o pieniądze, to ten budżet konsumuje proces administracyjny, czyli wszystkie kwestie związane z postępowaniem administracyjnym w trakcie prowadzenia tego procesu, jak również kolejne korzyści, które wynikają z procesu scaleniowego, czyli dokonanie różnego rodzaju zmian w dokumentach czy inwestycji na terenie gruntów, które obejmuje obszar scalenia.

Możemy tworzyć środowisko, które wspomaga. Natomiast scalenie wynika z wniosku złożonego przez zainteresowane strony, czyli 51% właścicieli, użytkowników gruntów, których ten obszar scaleniowy ma dotyczyć. Ta ustawa - warto to też podkreślić - dokonuje pewnej bardzo ważnej, istotnej zmiany. Chodzi o to, że to użytkownik tego gruntu, czyli rolnik, który np. prowadzi dzierżawę na jego terenie, może również znaleźć się w tej grupie 51% wnioskodawców, którzy wychodzą z inicjatywą wprowadzenia tego procesu w życie.

Otóż nie. To dotyczy tylko i wyłącznie tej ustawy i tylko tego procesu scaleniowego, czyli osoby dysponujące obszarem o powierzchni przynajmniej 1 ha, obszarem rolnym bądź leśnym, mogą brać udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym tego scalenia, natomiast nie mogą występować o jakieś dotacje czy jakiekolwiek inne korzyści, które przysługują rolnikom czy właścicielom gruntów rolnych. Były również pytania dotyczące tego, czy w wyniku tego postępowania jeden rolnik zostanie przesunięty, czy jego działki zostaną przesunięte z jednego miejsca na drugie, gminy czy powiatu. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Szanowni Państwo!

On także daje szansę na to, żeby ten proces prowadzić w sposób dynamiczny. My jako ministerstwo rolnictwa składaliśmy takie wnioski, inicjatywa z naszej strony miała miejsce, natomiast nie zyskało to aprobaty komisji czy Sejmu i skupiono się wtedy na innych - w opinii posłów czy części posłów być może ważniejszych - przepisach.

Wydaje mi się, że na wszystkie pytania, które tutaj padły, udzieliłem odpowiedzi. Również jesteśmy, oddajemy się do państwa dyspozycji, jeśli przyjdzie państwu do głowy jakieś inne pytanie, jakaś inna wątpliwość. Dziękuję, panie ministrze. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1344 i 1691) Bardzo proszę pana posła Grzegorza Lorka o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druki nr 1344 i 1691. Przypomnę, że projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie oraz doprecyzowanie funkcjonujących regulacji prawnych w Kodeksie cywilnym, mianowicie dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia na skutek wszczęcia mediacji lub złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, instytucji wyzysku, odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim posłankom i posłom za udział w pracach zarówno podkomisji, jak i komisji. Chciałbym tu też przekazać Izbie informację, że Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględniło postulaty społeczne i została wprowadzona poprawka, która ma na celu doregulowanie przedstawionych przez organizacje społeczne kwestii. No cóż, życie parlamentarne i Wysokiej Izby jest takie, że pewnie będziemy jeszcze raz nad tym procedować w komisji. Tak to już jest. Chcemy, żeby ten akt był, że tak powiem, najlepszy z możliwych i wszystkie siły polityczne się o to starają. W imieniu komisji wnoszę, aby Wysoki Sejm uchwalił załączony projekt ustawy. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Pierwszą osobą, która zabierze głos, będzie pan poseł - znany nam już - Grzegorz Lorek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druki nr 1344 i 1691. W projekcie przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie oraz doprecyzowanie funkcjonujących regulacji prawnych w Kodeksie cywilnym. Mianowicie są to: przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia mediacji lub złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, instytucja wyzysku, odpowiedzialność pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu i ostatnia kwestia, związana z art. 159 Kodeksu cywilnego, który w naszej ocenie stanowi wyłom przy wnoszeniu gruntów do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Wskazany przepis ma nikłe znaczenie praktyczne. Ponadto stosowanie zasad ogólnych oraz wymaganie aktu notarialnego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu takimi nieruchomościami. Należy zwrócić uwagę na to, że pojawiają się głosy, jakoby wierzyciele nadużywali tej instytucji, żeby osiągnąć przerwanie biegu terminu przedawnienia. Zatem w sytuacji gdy dojdzie do przerwania biegu terminu przedawnienia, termin ten liczy się od początku po ustaniu okoliczności, które uzasadniają jego zawieszenie. Natomiast w przypadku zawieszenia ten termin biegnie dalej od chwili, kiedy ustała przyczyna zawieszenia. Ustawa ma wyeliminować praktykę składania przez wierzycieli wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia. Pozwoli to na wyklarowanie sytuacji procesowej stron sporów oraz przywróci zawezwaniu do próby ugodowej jego pierwotny, właściwy cel, czyli zawarcie ugody. Z tego też względu klub Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje przedłożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druki nr 1344 i 1691, i wnosi o przyjęcie załączonego projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pani poseł Barbara Dolniak, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W tym przypadku będzie wprowadzone zawieszenie, a więc do tego terminu przedawnienia będzie się doliczać tylko i wyłącznie czas, na który nastąpiło zawieszenie jego biegu.

A więc trzeba będzie spełnić kilka przesłanek, by móc uchronić się od odpowiedzialności na podstawie tego przepisu. Projekt przewiduje również zmiany dotyczące art. 388 Kodeksu cywilnego. Przepis ten odnosi się do wyzysku. Zgodnie z projektem poszkodowany będzie teraz mógł według swojego wyboru żądać zmniejszenia swojego świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia albo unieważnienia umowy.

W tym przypadku trudno zgodzić się z takim rozwiązaniem. Jest ono niepotrzebne. Dotychczasowe brzmienie pozwala na szerokie rozumienie użytych w nim przesłanek.

W myśl słownika języka polskiego pojęcie „niedoświadczenie” oznacza również, że osoba niedoświadczona to osoba nieobeznana, łatwowierna, niewprawiona, nieporadna, niezorientowana czy nieznająca się. Również w orzecznictwie przesłanka niedoświadczenia odczytywana jest w kontekście określonego rodzaju stosunków prawnych jako brak doświadczenia w określonego rodzaju przedsięwzięciach.

Tym samym należy uznać ją za zbędną. Takie poszerzanie przepisów niczemu dobremu nie służy. To czyni ten przepis tylko bardziej skomplikowanym.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania odbędzie się, proszę państwa, kosztem daleko idącego ograniczenia swobody orzeczniczej sądów – a na tym powinno opierać orzekanie. To sądowi należy pozostawić ocenę, przy wzięciu pod uwagę konkretnych okoliczności sprawy, czy mamy do czynienia z rażącą dysproporcją świadczeń, czy też nie. Ponadto trzeba zauważyć, że wprowadzenie domniemania, że rażąca jest co najmniej dwukrotna dysproporcja świadczeń, w praktyce może ukształtować stanowisko, że nie są spełnione przesłanki wyzysku, jeżeli wartość świadczenia wyzyskanego przewyższa wartość świadczenia wzajemnego o 99% albo mniej. Należy również zauważyć, że w gospodarce rynkowej różnica cen niektórych produktów nie jest niczym nadzwyczajnym. W projekcie przewidziano, iż uprawnienia w nowelizowanym art. 388 § 1 wygasają z upływem 3 lat od dnia zawarcia umowy, a jeśli stroną jest konsument - z upływem aż 6 lat. Składamy poprawkę, w której przewiduje się, że w miejsce 2-letniego terminu dla wszystkich będzie termin 3-letni. Konsument może skorzystać (Dzwonek) z innych rozwiązań, np. z art. 385 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli klauzul abuzywnych. Przysługują mu również inne świadczenia i możliwości wynikające z prawa konsumenckiego czy nawet z art. 58 Kodeksu cywilnego. Jest to bardzo duże wydłużenie, niczym nieuzasadnione. Pamiętam, że w poprzedniej kadencji PiS, wnosząc zmiany dotyczące terminów przedawnienia, skracał je i gdy wskazywałam, że będą dotyczyć również konsumentów, przyjmował to do wiadomości, a teraz w sposób niczym nieuzasadniony, bo nie wynika to z żadnej analizy projektu ustawy, wydłuża ten termin do aż 6 lat, proszę państwa, z 2 lat, które obowiązują w tej chwili zgodnie z przepisem. Tym samym składamy poprawki do tego projektu ustawy, licząc, że będą one przedmiotem merytorycznej dyskusji - bo taka dyskusja, a nie polityczna, powinna się odbywać w nadzwyczajnej komisji kodyfikacyjnej, gdzie tworzymy przepisy stanowiące bazę, podstawę funkcjonowania systemu prawnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. Tak trochę z racji tego, że jesteśmy z Zagłębia, minutę pani dodałem. Pani posłanka Katarzyna Ueberhan, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, zawartego w druku nr 1344, wraz ze sprawozdaniem komisji, zawartym w druku nr 1691. Główne zmiany wprowadzone niniejszym przedłożeniem zakładają przede wszystkim łatwiejsze podważenie nieuczciwych umów, trudniejsze przerwanie biegu przedawnienia przez wierzyciela, jak też brak odpowiedzialności osób niesamodzielnych, a wspólnie zamieszkujących z rodzicami - nie będą już odpowiadać za długi czynszowe swoich rodziców. Zmiany dotyczące przepisów o wyzysku to reakcja na nieuczciwe praktyki rynkowe w postaci zawierania umów o skutkach analogicznych właśnie do wyzysku, lecz formalnie niemieszczących się w zakresie stosowania obecnie obowiązującego art. 388 Kodeksu cywilnego. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju sprzedaż garnków, pościeli czy innych artykułów wyposażenia domowego o rzekomo nadzwyczajnych parametrach, podczas gdy ich jedyną wyjątkową cechą była zazwyczaj nadzwyczaj wysoka cena. Podobnie w tym samym katalogu nieuczciwych praktyk zawiera się oferowanie osobom w trudnej sytuacji życiowej, postawionych pod tzw. przysłowiową ścianą, stosunkowo niskich pożyczek na wysoki procent, i to pod zastaw już o wiele więcej wartych nieruchomości. Analogiczne nieuczciwe praktyki spotykamy też w niektórych umowach franczyzowych, w których charakter wzajemnych zobowiązań daleki jest od wzajemnej równowagi. Niniejsze przedłożenie to próba rozwiązania tego typu problemów i swego rodzaju koło ratunkowe dla ofiar oszustów. W sytuacjach takich jak te wymienione powyżej słabość strony wyzyskanej nie polega na niedołęstwie czy niedoświadczeniu, o których mowa obecnie w art. 388 Kodeksu cywilnego, lecz na braku wiedzy co do faktycznych skutków zawieranej umowy. Projekt przewiduje rozszerzenie przesłanek wyzysku o wykorzystanie braku dostatecznego rozeznania.

Poza tym obecnie można dochodzić tylko zmniejszenia świadczenia lub zwiększenia świadczenia drugiej strony, a tylko w sytuacji gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione - unieważnienia umowy. Teraz to od pokrzywdzonej strony będzie zależało, które z tych trzech rozwiązań wybierze. Kolejnym z rozwiązań w proponowanym przedłożeniu jest zawieszenie biegu przedawnienia przy mediacjach i rozmowach o ugodzie w związku z dotychczasowym nadużywaniem przez wierzycieli instytucji zawezwania do próby ugodowej i praktyką składania przez wierzycieli wniosku o zawezwaniu do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia. Czy proponowane rozwiązanie faktycznie wyeliminuje ten proceder i skutecznie ograniczy liczbę spraw wpływających do sądu z tego tytułu, jak zakładają projektodawcy? Mam nadzieję, że tak. Kolejne rozwiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego pełnoletnie osoby wspólnie zamieszkujące z najemcą nie będą już ponosić faktycznej odpowiedzialności za czynsz i inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. W toku prac komisji oraz podkomisji zgłaszano wiele wątpliwości i poprawki, w tym poprawkę społeczną, którą uwzględniono. Po uwzględnieniu poprawek zgłaszanych w toku prac komisji oraz przy drugim czytaniu, korygujących wątpliwości co do niektórych szczegółowych rozwiązań, mając na uwadze, że projektowane zmiany są oczekiwane i potrzebne oraz pomimo wszystko wpływają na poprawę sytuacji podmiotów znajdujących się na słabszej pozycji w dochodzeniu swoich praw, klub Lewicy poprze niniejsze przedłożenie. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Faktycznie podejmujemy wspólnie próbę nowelizacji Kodeksu cywilnego i procedury cywilnej, działając w bardzo słusznym legislacyjnym kierunku wyjścia naprzeciw osobom, które w dotychczasowym porządku prawnym bardzo łatwo mogły paść ofiarą różnych nieuczciwych praktyk. Wszyscy dobrze znamy powszechny proceder zapraszania osób starszych, osób, które nie do końca są w stanie rozeznać, jak prezentują się oferty sprzedaży słynnych garnków, różnych innych produktów oferowanych po częstokroć bardzo, bardzo znacząco zawyżonych cenach.

Bardzo często tak bywało, dlatego my jako klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego z uznaniem podchodzimy do tego projektu.

Myślę, że poprawki, jak również postulaty prezentowane chociażby przez Radę Przedsiębiorczości, też powinny zyskać uznanie w toku dalszych prac.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, drogi Michale. Proszę bardzo. Czcigodny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Niestety wspólnym mianownikiem takich transakcji jest przede wszystkim wysoka cena nabywanych produktów, ponadto bardzo niekorzystne warunki wyjścia z tego typu umów. To jest problem moralny, społeczny i prawny, bo seniorzy często bywają po prostu bezbronni wobec takich nowoczesnych technik sprzedażowych. Często i słusznie zwracają się później z prośbą o pomoc do państwa. Odpowiedzią na wyzwanie jest oczywiście modyfikacja treści słynnego art. 388 k.c. i z satysfakcją przyjmujemy pojawienie się dodatkowej przesłanki braku dostatecznego rozeznania.

Zdecydowanie ułatwi do zdefiniowanie tzw. wyzysku.

Doceniamy i popieramy prokliencki i prokonsumencki charakter tych przepisów. Ono idzie z duchem czasu. W prawie cywilnym również pod wpływem prawa europejskiego wprowadza się przepisy, które chronią słabszą stronę umowy. Wydaje się, że jedyną w pewien sposób pokrzywdzoną grupą społeczną będą studenci 2. roku prawa, którzy zjawisko wyzysku będą musieli definiować na egzaminach, a ono będzie dużo bardziej skomplikowane niż w obecnym stanie prawnym. Ale to jest mała cena za te dobre przepisy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, dziewięć osób zapisało się do pytań. Zamykam listę. Proszę pana posła Rafała Adamczyka z klubu parlamentarnego Lewica o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Tutaj czytamy, że projekt ustawy dotyczy wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu usprawnienie i doprecyzowanie funkcjonujących regulacji prawnych.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Zapis w swoich intencjach uznaję za właściwy i potrzebny, ale czy nie pozostaje on w sprzeczności z innymi przepisami? Otóż osoba obarczona współodpowiedzialnością finansową za zobowiązania czynszowe powinna posiadać określone prawa, których nie gwarantuje jej system prawny. Osoba zamieszkująca we wspólnym lokalu z najemcą głównym nie ma żadnych praw do kontroli stanu zadłużenia, nie ma też żadnych formalnych praw do występowania jako strona w ewentualnych sporach czy negocjacjach. Jest to forma ubezwłasnowolnienia finansowego. Czy projekt nie nakłada na obywateli obowiązku spłaty zadłużenia, którego te osoby nie są świadome? Dziękuję bardzo. Pan poseł Zdzisław Wolski, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo!

Uważam, że użyte w projektowanym projekcie słowo „rozeznanie” jest zbyt ogólne i szerokie, a w szczególności nie jest doprecyzowane, czego dotyczy brak rozeznania. Nieprecyzyjny i subiektywny charakter rozeznania czy szczególnie braku rozeznania utrudni dowodzenie tego w procesie sądowym. Będzie to trudne do zweryfikowania przez biegłych sądowych i będzie to dawało pole do nadużyć dłużnikom, a czasami wierzycielom.

Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proponowany pkt 6 w art. 121 określa, że bieg roszczeń objętych wnioskiem o próbę ugodową ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania pojednawczego. Budzi to pewną wątpliwość. Zakładając, że bieg przedawnienia roszczenia zakończyłby się w czasie postępowania pojednawczego będącego w toku, można przyjąć, że przedawnienie nastąpi z chwilą zakończenia postępowania objętego wnioskiem o wezwanie do próby ugodowej.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby na wyeliminowanie nadużyć procesowych związanych ze składaniem kolejnych wniosków o zawieszenie w związku z podjęciem próby ugodowej z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu wierzyciela. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku!

Gdyby to dotyczyło polityków, to myślę, że w kontekście szalejącej drożyzny, inflacji zarówno pan premier Morawiecki, jak i prezes Banku Centralnego pan Glapiński byliby właśnie odbiorcami tego typu oświadczeń. Natomiast moje pytanie dotyczy art. 688 i bardzo bym prosił o odpowiedź. Czy spółdzielnie mieszkaniowe będą miały jakieś narzędzia do tego, żeby ten przepis, który wprowadza solidarną odpowiedzialność za zobowiązania, mogły stosować w praktyce? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponowane zmiany zakładają m.in., że zawezwanie do próby ugodowej stanie się czynnością procesową zawsze wpływającą na bieg przedawnienia, powodującą zawieszenie tego biegu bez względu na cel, w jakim zostało dokonane. Z jednej strony zatem chcecie wyeliminować pozorność składania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jako narzędzia wykorzystywanego do wydłużania terminu przedawnienia roszczenia, a z drugiej strony wyłączacie stosowany w praktyce sądów wymóg badania celu składania takiego wniosku. Nie bardzo rozumiem, do czego w takim razie tak naprawdę zmierzamy. Przecież dokonana w taki sposób zmiana przepisów będzie tylko pozorem i nie przyniesie żadnej korzyści, i pogłębi już i tak panujący za waszych rządów (Dzwonek) chaos w sądach. Dziękuję. Pan poseł Andrzej Szejna, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! W obecnym stanie prawnym art. 388 k.c. stanowi, iż umowa jest wadliwa, gdy spełnione zostaną przesłanki natury obiektywnej i subiektywnej. Przesłanka obiektywna znajduje wyraz w kwalifikowanej dysproporcji świadczeń stron.

Przedłożony projekt ustawy dodaje w tym katalogu także brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy. Zgodnie z projektowanym przepisem, jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, domniemywa się, że niewspółmierność świadczenia ma charakter rażący.

Dziękuję. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Trzeba pamiętać, że zbyt długi termin niesie za sobą ryzyko zmiany wartości świadczeń, w tym także na niekorzyść wyzyskanego, w związku z czym, wprowadzając termin, nie można tego czynić dowolnie (Dzwonek), decydować się na cokolwiek. Trzeba rozważać w każdym przypadku interes obu stron. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pani minister Katarzyna Frydrych odpowie na państwa pytania. Zapraszam, pani minister.

Wysoka Izbo! W pierwszej kolejności pragnę złożyć wyrazy podziękowania za wkład Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach pod przewodnictwem pana posła Piotra Saka oraz podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego na czele z przewodniczącym panem posłem Grzegorzem Lorkiem w pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Nie zauważyłam, żeby w trakcie prac zarówno podkomisji, jak i komisji toczyła się jakakolwiek dyskusja polityczna. Moim zdaniem była to dyskusja bardzo merytoryczna. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

Dookreślenie przesłanek wyzysku, jakim są niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania, doprowadzi do sprecyzowania, że obie te okoliczności mają się odnosić wyłącznie bezpośrednio do przedmiotu umowy.

Strona rządowa jest przekonana, że projekt w brzmieniu ze sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach nie będzie budził problemu w zakresie stosowania prawa, jak również stanowi odzwierciedlenie potrzeb społeczeństwa w odniesieniu do potrzeb ochrony ich praw i interesów. Odniosę się teraz do pytań, które zostały zadane w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Po pierwsze, chciałabym zwrócić uwagę - odpowiadam na pytanie pana posła Rafała Adamczyka - że nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że przeciwko wprowadzeniu projektowanej regulacji świadczyć miałby fakt, że właściciel, w przypadku gdy nieruchomość jest w posiadaniu osoby, której tytuł prawny do gruntu opiera się na decyzji administracyjnej, nie ma innej możliwości zapobieżenia terminowi przed doprowadzeniem do unieważnienia wszystkich wydanych dotąd decyzji niż poprzez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Taki argument jest właśnie akademickim przykładem wykorzystywania instytucji zawezwania sprzecznie z jej celem zamiast zawarcia ugody. Chodzi bowiem wnioskującemu o przerwanie biegu terminu zasiedzenia, a przecież nie temu ma służyć postępowanie pojednawcze. Należy wskazać, że zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2020 r. czynność przed organem administracyjnym zmierzająca do uchylenia decyzji np. wywłaszczeniowej stanowi taką manifestację, a co za tym idzie - skutkuje przerwaniem biegu terminu zasiedzenia. Innego typu czynnością jest natomiast przykładowe wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości czy też uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Nie ma zatem tutaj zagrożenia, że eliminacja skutków w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej doprowadzi do jakichś systemowych niekonsekwencji i perturbacji związanych z biegiem terminu zasiedzenia.

Tak naprawdę chodziło o to, aby osiągnąć cel, który jest tożsamy z tym, który mamy aktualnie, jeśli chodzi o brzmienie art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który prowadzi do zwolnienia od odpowiedzialności za zobowiązania czynszowe pełnoletnich wstępnych z przyczyn, które istnieją obiektywnie. Jeśli chodzi o przesłankę braku rozeznania, która pojawiła się jako nowa przesłanka w art. 388, to należy stwierdzić, że z obserwacji wynika, że słabość strony wyzyskanej często polega nie tylko na jej niedołęstwie czy niedoświadczeniu, lecz także na braku świadomości co do faktycznych skutków zawieranej umowy bądź wiedzy specjalistycznej pozwalającej na ich ustalenie. Wprowadzenie przesłanki braku dostatecznego rozeznania nie wiąże się z całkowitym zwolnieniem z konieczności dokonania choćby wstępnej orientacji czy oceny co do przedmiotu umowy, jednak to na oferencie spoczywa obowiązek przedstawienia drugiej stronie wszelkich informacji, które dotyczą przedmiotu umowy, praw, obowiązków wynikających z umowy, co ma umożliwić kontrahentowi świadome podjęcie decyzji. W naszej ocenie brak doświadczenia nie jest równoznaczne z tą nową przesłanką dotyczącą braku dostatecznego rozeznania. Już odnosiłam się do kwestii art. 688, mówiąc, że nie jest to nowa regulacja. Podobną regulację mamy również w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeśli natomiast chodzi o kwestię związaną z tym, że nakładamy na sądy obowiązek badania celu złożenia wniosku, to absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. Takiego obowiązku sąd nie ma.

Tym samym nie jest prawdą, aby był ten cel badany, jeśli chodzi o złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Jeśli chodzi o termin, który został wydłużony - to jest termin zawity, przewidziany w art. 388 Kodeksu cywilnego - to w naszej ocenie wydłużenie tego terminu ma na celu danie gwarancji osobie, która w momencie zawarcia umowy była niedoświadczona, znajdowała się w przymusowym położeniu lub nie posiadała dostatecznego rozeznania. Chcę zauważyć, że jest to termin, który nie liczy się od dnia wymagalności roszczeń, ale od dnia zawarcia umowy. W naszej ocenie utrzymanie dotychczasowego, krótkiego terminu zawitego ze względów aksjologicznych jest niepożądane, tym bardziej że ta osoba może zorientować się dużo później niż w czasie 2 lat od dnia zawarcia umowy, że tak naprawdę padła ofiarą wyzysku, a przecież chodzi o to, żeby chronić obywateli najsłabszych. Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Fabisiak, to nie wiem, czy je zrozumiałam dobrze. Jeśli je zrozumiałam błędnie, to udzielimy odpowiedzi na piśmie. Ale chciałam zaznaczyć, po pierwsze, kwestię następującą: jeśli to pytanie dotyczyło zobowiązań za długi spadkowe, to ta regulacja nie dotyczy tej kwestii. Natomiast jeśli dotyczyło kwestii związanej z odpowiedzialnością pełnoletnich zstępnych, to w mojej ocenie ta odpowiedzialność jest tylko i wyłącznie za okres, kiedy pełnoletni zstępni stale zamieszkują z najemcą. Innej odpowiedzialności ten przepis nie przewiduje.

Chodzi o pełnoletnich zstępnych stale zamieszkujących z najemcą przez ten okres, którego dotyczą powstałe zobowiązania.

Chodzi o sytuację, kiedy osoba jest zameldowana, ale nie mieszka w domu, bo została z tego domu wypędzona. Jest zameldowana, w związku z czym samorząd uznaje ją za osobę mieszkającą. Czasami można udowodnić, że nie zamieszkiwała, ale nie zawsze. Taka osoba w pełni odpowiada za zadłużenia czynszowe i musi je spłacać, a samorząd nie ma podstawy prawnej, aby umorzyć to zadłużenie na rzecz tej osoby. Nawet jeśli właściciel nie zamieszkuje. Ale jest poważniejsza sprawa: wówczas na ogół nie są podpisywane umowy z młodą osobą, która pozostaje bez dachu nad głową. Bardzo proszę, pani minister. Panie Marszałku! Wydaje mi się, że to jest zawsze, pani poseł, kwestia dowodowa. To sąd musi zbadać, czy zaistniała przesłanka zamieszkiwania, bo czym innym jest zameldowanie, a czym innym jest faktyczne zamieszkiwanie w tym lokalu. Trzeba to rozróżnić. Fakt, że ktoś jest zameldowany w lokalu, nie oznacza, że w nim po prostu przebywa i zamieszkuje.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, na podstawie art. 95 ust. 2 regulaminu Sejmu kieruję ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu przedstawienia sprawozdania. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana ministra Macieja Miłkowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło przedstawić państwu projekt ustawy o wyrobach medycznych.

Oba te akty wspólnotowe mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, przyjmując jako podstawę wysoki poziom ochrony zdrowia, z myślą o pacjentach, użytkownikach, z uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców działających w tym sektorze. W szczególności ta ustawa określa właściwość poszczególnych organów w tym zakresie, obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, zasady prowadzenia reklamy, system kar administracyjnych. Celem tej ustawy jest wprowadzenie i uregulowanie kwestii, które są możliwe do uregulowania, które ww. rozporządzenia pozostawiają do decyzji państw członkowskich, oraz stworzenie ram prawnych dla właściwej i skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków właściwych organów i podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na terytorium naszego kraju. W kompetencji naszego kraju i wszystkim krajów pozostawiono możliwość uszczegółowienia zasad sprawowania nadzoru nad podmiotami prowadzącymi obrót wyrobami medycznymi na terytorium RP, wprowadzenia przepisów regulujących możliwość regenerowania i dalszego używania wyrobów medycznych jednorazowego użytku, żądania od producentów wyrobów medycznych na zamówienie wykazu wyrobów, które zostały udostępnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji udziału komisji etycznych w ocenie badania klinicznego, tego, w jaki sposób prezes urzędu nadzoruje badania kliniczne wyrobów medycznych, ustalania informacji szczegółowych dotyczących tego, w jaki sposób mają być oznakowane wyroby medyczne, w jakich językach mają być określone.

Wyrażam zgodę.

Zapraszam, panie prezesie. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Na wstępie dziękuję panu ministrowi za kompleksowe przedstawienie projektu ustawy, który dla mnie jako przedstawiciela centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawie wyrobów medycznych ma istotne znaczenie. Projektowane przepisy będą służyć przede wszystkim skutecznemu stosowaniu rozporządzeń, które wymienił pan minister, czyli 745 i 746 Parlamentu Europejskiego i Rady. Akty te mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze tych wyrobów. Prezes urzędu został wyznaczony jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach związanych z wdrażaniem przepisów unijnych rozporządzeń oraz organ odpowiedzialny za jednostki notyfikowane, które certyfikują wyroby medyczne. Jest to nowe zadanie w stosunku do już posiadanych kompetencji i realizowanych w oparciu o przepisy dotychczasowej ustawy. Warte podkreślenia z punktu widzenia właściwej realizacji nowych zadań jest wyposażenie prezesa urzędu w uprawnienie do żądania udostępnienia mu przez organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne administracji publicznej wszelkich posiadanych informacji dotyczących obrotu wyrobem, systemem lub zestawem zabiegowym. Projekt zakłada, że prezes urzędu będzie organem uprawnionym do dokonywania w drodze decyzji administracyjnych klasyfikacji wyrobów w przypadku sporu pomiędzy producentem a jednostką notyfikowaną, która certyfikuje wyroby medyczne, tak jak wspomniałem, co do klasy ryzyka, w jakiej powinien znaleźć się dany wyrób medyczny. Mając na względzie wyzwania, jakie postawiła przed nami epidemia COVID-19, wskazać należy na istotną regulację, w przypadku której prezes urzędu na należycie uzasadniony wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, konsultanta krajowego, konsultanta wojewódzkiego, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub prezesa NFZ będzie mógł wydawać, w drodze decyzji administracyjnej, pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonego wyrobu, w przypadku którego nie przeprowadzono procedur oceny zgodności, ale którego używanie leży w interesie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia pacjentów. Nie bez znaczenia jest, iż przy wykonywaniu zadań wynikających z rozporządzeń nr 745 i 746 prezes urzędu współpracuje i wymienia informacje z właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej. Harmonizacja działań i współpraca międzynarodowa ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów medycznych, który jest bez wątpienia ogromnym rynkiem wyzwań, ale także możliwości. Dodatkowo celem projektowanej ustawy jest uregulowanie kwestii pozostawionych przez rozporządzenia do decyzji państw członkowskich i ich rozstrzygnięcia na poziomie wyłącznie krajowym. W związku z tym prezes będzie sprawował również nadzór nad reklamą wyrobów medycznych dotychczas nigdzie nieuregulowaną w przepisach prawa. Projekt zakłada zastąpienie obecnych przepisów karnych pieniężnymi karami administracyjnymi, co niewątpliwie pozwoli na efektywniejszy nadzór i sprawniejsze sankcjonowanie nagannych zachowań. Należy pamiętać, że zapewnienie wykonania przepisów rozporządzeń i ustawy poprzez ustanowienie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji za ich naruszenie jest jednym z podstawowych celów omawianych regulacji. W przedmiotowym zakresie prezes urzędu będzie wydawał decyzje administracyjne. W projekcie przewidziane jest także wprowadzenie przepisu uprawniającego organ do odstąpienia od wymierzania kar pieniężnych, jeżeli zdarzenie miało charakter incydentalny, nie stwarzało ryzyka, a podmiot, najpóźniej w terminie wskazanym przez prezesa urzędu, ministra właściwego do spraw zdrowia albo głównego inspektora sanitarnego, przy prowadzeniu czynności, w trakcie których stwierdzono uchybienie prawa, podjął działania w celu ich usunięcia i poinformował właściwy organ o ich podjęciu. Mając na względzie to krótkie podsumowanie, pokładam nadzieje, że kompleksowe stosowanie przepisów ustawy i rozporządzeń unijnych pozwoli na utrzymanie wysokich norm jakości i bezpieczeństwa w przypadku wyrobów medycznych oraz harmonizację zasad wprowadzania ich do obrotu i używania na rynku unijnym, przede wszystkim zaś zagwarantuje szerszą identyfikację wyrobów medycznych i ich producentów, a także innych podmiotów w łańcuchu dostaw, zapewniając tym samym skuteczny nadzór, a użytkownikom - łatwiejszy dostęp do informacji na temat tych wyrobów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Barbara Dziuk. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość chcę przedłożyć informację oraz stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych, druk nr 1764. Celem przedstawionego projektu ustawy o wyrobach medycznych jest dostosowanie polskiego prawa do rozporządzeń Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania rynku wyrobów medycznych i zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia naszego społeczeństwa. Uporządkowanie dotyczy działalności wszystkich firm działających w sektorze medycznym. W ustawie określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie przekazywanych informacji na temat obrotu tymi wyrobami. Projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń Unii Europejskiej, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku dotyczące wyrobów medycznych. Chodzi o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem działalności małych i średnich firm w tym sektorze. W szczególności określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych. Najważniejsze rozwiązania proponowane w ustawie dotyczą tego, że prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie wydawał decyzje administracyjne w sytuacjach określonych przez przepisy Unii Europejskiej. Prezes urzędu będzie mógł żądać informacji o wyrobach medycznych m.in. od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów prowadzących taki obrót bądź stosujących te wyroby. Dotyczyć to będzie także wykazu wyrobów medycznych na zamówienie, które zostały udostępnione na terytorium Polski, jak również producenta wyrobu wykonanego na zamówienie. Wprowadzono obowiązek przekazywania m.in. deklaracji zgodności, instrukcji używania oraz oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu albo przekazywanych do oceny działania lub stosowanych na terytorium Polski.

Określono zasady regeneracji wyrobów medycznych jednorazowego użytku, wprowadzając zakaz używania w Polsce zregenerowanych wyrobów jednorazowego użytku. Wprowadzono również system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Dariusz Klimczak w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Oceniając całokształt planowanej ustawy, można powiedzieć, że jej celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w ochronie zdrowia, że została stworzona z myślą o pacjentach i użytkownikach korzystających z określonych wyrobów medycznych. Implementacja odpowiednich przepisów europejskich ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. W oczywisty sposób niniejsze przepisy będą dotyczyć przedsiębiorców działających w tym sektorze.

Objęte nadzorem mają zostać liczne grupy wyrobów wymienionych w załączniku XVI do rozporządzenia. Chodzi np. o soczewki kontaktowe, substancje przeznaczone do stosowania przy wypełnianiu skóry twarzy, sprzęt do liposukcji czy lasery do usuwania tatuaży lub włosów.

Wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów, ale nie przeszkodzi przedsiębiorcom. Dziękuję bardzo. Stanowisko Koalicji Obywatelskiej przedstawi pan poseł Rajmund Miller. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej - Platformy Obywatelskiej wobec rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych, druk nr 1764.

Projekt dotyczy funkcjonowania rynku wyrobów medycznych w Polsce. Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia przez zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie obrotu wyrobami medycznymi i wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Zawiera również szczegółowe zapisy dotyczące zadań w wymienionym obszarze, które są dedykowane Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz obowiązki w zakresie przekazywania określonych w ustawie informacji przez podmioty gospodarcze, o czym przed chwilą mówił pan prezes.

Zostaje wprowadzony obowiązek przekazywania m.in. deklaracji zgodności, instrukcji używania, oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu, przekazanych do oceny działania lub stosowanych na terytorium Polski. Wprowadzone zostają zasady regeneracji wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Szanowni Państwo!

Po pierwsze, likwidacja obowiązku informowania prezesa urzędu o wyrobach sprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej przez dystrybutorów i inne podmioty, które nie przekazują danych do europejskiej bazy danych.

Uwag jest bardzo dużo. Uważamy, że cel projektu jest słuszny. Myślę, że w trakcie obrad komisji okaże się, jakie są szczegółowe zapisy tego projektu.

Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Marek Rutka w imieniu klubu Lewica. Zapraszam. Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ustawy o wyrobach medycznych ma służyć stosowaniu dyrektywy i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Nadrzędnym celem tych regulacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której na terenie Wspólnoty zagwarantowany zostanie jednorodny i możliwie najwyższy poziom ochrony zdrowia, ukierunkowany na pacjentów, to jest szczególnie ważne, a także uwzględniający interesy małych i średnich przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Z uwagi na to, że wyroby medyczne są bardzo szczególnymi produktami, ryzyko związane z ich użytkowaniem może mieć bardzo poważne konsekwencje w przyszłości dla pacjentów czy użytkowników. Stąd też celowe jest wprowadzenie regulacji w tym obszarze. Jest to instytucja z ponad 20-letnią tradycją i to jest na pewno dobre rozwiązanie, że nie tworzy się nowego organizmu. Zgodnie z założeniami pozwoli to na efektywniejszy nadzór sprawowany przez prezesa urzędu oraz skrócenie postępowań w sprawie nakładania kar. Z zadowoleniem należy przyjąć, że w projekcie przewidziano również wprowadzenie przepisu uprawniającego organ do odstąpienia od wymierzenia kar pieniężnych, jeśli zdarzenie miało charakter incydentalny, nie stwarzało ryzyka, a podmiot, który podjął działania w celu ich usunięcia, poinformował właściwy organ o ich podjęciu. Przepis ten ma na celu uniknięcie sytuacji, w których przedsiębiorcy lub inne podmioty będą karani, gdy naruszenie przepisu będzie miało jedynie charakter incydentalny. Projekt przewiduje udostępnianie informacji o podmiotach i osobach sprzedających wysyłkowo wyroby w sytuacji, w której prezes urzędu nie posiada informacji umożliwiających mu wykonywanie obowiązków nadzorczych. Biorąc pod uwagę szereg patologii, do których dochodzi w przypadku sprzedaży wysyłkowej produktów medycznych, uchodzących za medyczne i paramedyczne, jak chociażby syntetyczne kołdry z lamy, magiczne poduszki przywracające władzę w kończynach czy mikstury eliminujące syndrom niespokojnych stóp, wprowadzenie nadzoru nad sprzedażą wysyłkową jest kierunkiem słusznym i trzeba mieć nadzieję, że przynajmniej częściowo ograniczy wysokodochodowe szarlataństwo.

W projektowanych przepisach zmieniających ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza się również wymóg, aby pacjentom, którym wszczepiono dany wyrób medyczny, udostępniano wraz z tą, można powiedzieć, usługą, wraz z kartą implantu wszelkie stosowne informacje przekazywane przez producenta wyrobu i pozwalające na identyfikację wyrobu. Wyrób przeznaczony do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej ma mieć tzw. interfejs użytkownika w języku polskim lub w postaci zharmonizowanych. W przypadku wyrobów sterowanych lub komunikujących się z użytkownikiem za pomocą komend głosowych interfejs oraz komendy muszą być w języku polskim.

Aby to było jednoznaczne, to dobrze, że zostanie wprowadzony nakaz, aby te urządzenia komunikowały się z pacjentem w języku polskim. Przepisy mają również określać pewne zakazy i ograniczenia dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Z naszego punktu widzenia klub Lewicy na pewno nie jest do końca zadowolony z tych regulacji, które tutaj są proponowane, stąd też w zakresie wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby przedstawimy stosowne poprawki. Kolejne zastrzeżenie dotyczy braku regulacji odnośnie do zaprzestania publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy oraz publikacji wydanej decyzji w miejscach lub w środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama. To znaczy, jeśli reklama wprowadza w błąd potencjalnych pacjentów, powinna być w trybie administracyjnym usunięta.

Pan poseł Wojciech Maksymowicz w imieniu koła Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rządowy projekt jest wynikiem konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania rynku wyrobów medycznych. Przepisy unijne wprowadziły wiele elementów regulacyjnych, które mają na celu bezpieczeństwo użytkowania tych wyrobów. Rozwój badań wdrożeniowych i technologii wymaga takiego podejścia, ograniczając jednak wiele wcześniejszych, bardziej wolnościowych zasad. W projekcie zwiększa się kompetencje prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Swoją drogą jest to literacko straszna nazwa, którą można by przy okazji procesu legislacyjnego spokojnie skrócić.

Dookreślono obowiązki komisji bioetycznych i zakończono możliwości regeneracji wyrobów jednorazowych.

Ale już jesteśmy na poziomie partnerskim w Unii Europejskiej i trzeba to zaakceptować.

Nie mamy wątpliwości, że projekt powinien być dopuszczony do dalszego procedowania. Dziękuję. Wyznaczam czas - 1 minuta. Bardzo proszę, pani poseł. Oczywiście, że tak. Pierwsze pytanie zada pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Projekt dotyczy zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych dla diagnostyki in vitro. Jako podstawę przyjęto wysoki poziom ochrony zdrowia z myślą o pacjentach i użytkownikach. Panie ministrze, programy finansowania zabiegów in vitro kosztują i zapewne pan o tym doskonale wie. Czy planują państwo rozszerzyć programy wsparcia Polek i Polaków o wsparcie finansowe par chcących mieć potomstwo? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze!

Wykorzystuje ona, powiedziałbym, naturalną skłonność wszystkich rodziców do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo i dobrostan swojemu potomstwu.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Teraz, w okresie pandemii zakupy przez Internet powinny być codziennością, a dla osób z niepełnosprawnością na pewno są zdecydowanie bezpieczniejsze. Obecne przepisy pozwalają na refundację zakupu przez Internet wyrobów medycznych, które kupują co miesiąc, np. cewników, sprzętu stomijnego. A co z wyrobami, sprzętem medycznym, które osoby z niepełnosprawnością kupują rzadziej? Dlaczego w takiej sytuacji refundacja nie jest możliwa? Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Art. 5 projektu zakłada przekazywanie prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych imion, nazwisk, numerów PESEL, adresów zamieszkania, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej osób uczestniczących w obrocie wyrobami, systemem lub zestawami zabiegowymi określonymi w projekcie. Do jakich celów wspomniany urząd potrzebuje adresów zamieszkania tych osób i w jaki sposób te dane będą one przetwarzane? Czy zewidencjonowana osoba będzie mogła żądać usunięcia swoich danych z ewidencji urzędu, co gwarantują nam przepisy RODO? Moje pytanie do pana ministra, poproszę o odpowiedź na piśmie, dotyczy niezgodności omawianego projektu z obowiązującą w naszym kraju dyrektywą Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, która w precyzyjny sposób określa wszystkie jednostki administracyjne (Dzwonek) mające prawo do wglądu w dane osobowe oraz ich przechowywanie i przetwarzanie. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED zwróciła uwagę na przewidziane w obecnym projekcie wielomilionowe kary dla dystrybutorów wyrobów medycznych za błędy formalne w oznakowaniu wyrobów. Izba w opublikowanym stanowisku wyraża obawy, iż poziom tych kar obniża atrakcyjność produkowania wyrobów medycznych w Polsce i konsekwentnie sprawi, że te firmy wycofają się z produkcji w Polsce. Kary są nawet pięćdziesięciokrotnie wyższe niż w przypadku przepisów dotyczących leków czy żywności oraz znacznie wyższe niż analogiczne kary w innych krajach Unii Europejskiej. Sprzeciw wobec tych zapisów w stanowisku przekazanym do Sejmu wyraziło 15 organizacji, m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali itd. Panie ministrze, dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie aż tak wysokich kar? Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra o część dotyczącą zakazu reklamy. Chodzi o wprowadzenie dodatkowego zakazu reklamy wyrobów przeznaczonych do używania przez osoby posiadające określone kwalifikacje. Nie ma tam konkretnego wyjaśnienia, o jakie wyroby chodzi, ale w szczególności nie ma tego, jakie kryteria ma spełniać osoba posiadające określone kwalifikacje.

Ale to powinno być precyzyjnie uregulowane, tym bardziej że może dojść do wymierzania wysokich, a czasami bardzo wysokich kar. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Trwająca pandemia sprawiła, że zapotrzebowanie na wyroby medyczne znacząco wzrosło i niejako wymusiło zmianę przepisów w tym obszarze. Jednak, gdyby nie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, nawet byście nie zaczęli dyskusji na ten temat. Wasz projekt ustawy o wyrobach medycznych przewiduje wysokie kary administracyjne dla podmiotów, które nie zastosują się do nowych regulacji. Katalog tych sankcji, ich zakres i wysokość są w niektórych przypadkach nieproporcjonalne do rodzaju przewinienia i wielkości firmy. Proszę o odpowiedź na pytanie, skąd pewność, że przepisy nie będą powodować obaw np. o ich niesłuszne nakładanie, czego efektem mogą być przeniesienia firm za granicę i ucieczki potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji utrudnienia (Dzwonek) dla pacjentów do dostępnych na rynku wyrobów medycznych. Pani poseł Iwona Hartwich, Koalicja Obywatelska. Nie ma. Pan poseł Maciej Kopiec, klub Lewica. Wysoka Izbo! Dlaczego Sejm może rozdawać długopisy reklamowe opatrzone swoim logo, natomiast przedstawiciele handlowi branży medycznej nie będą mogli tego robić? Projektowane przepisy dotyczące wyrobów medycznych nie poruszają w ogóle tematu reklamy stanowiącej przypomnienie pełnej reklamy oraz nie regulują katalogu dozwolonych przedmiotów opatrzonych znakiem reklamującym dany wyrób medyczny. Efekt jest taki, że firmom łatwiej będzie wręczyć czajnik elektryczny z zamieszczonymi wszystkimi informacjami niż zwykły długopis. Ministerstwo Zdrowia chce zmniejszenia kolejek do lekarzy, jednak wizja darmowego czajnika zamiast długopisu może zwiększyć kolejki w przychodniach. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Jak wiemy, ten projekt ustawy to dostosowanie do prawa unijnego naszego prawa krajowego. Mówimy tutaj o reklamie i mam krótkie, jasne pytanie: Jakie zasady reklamy wyrobów medycznych będą obowiązywały po wprowadzeniu tej ustawy? Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Wprowadzacie państwo rozwiązanie i nadzór prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nad określonymi wyspecyfikowanymi zadaniami, które są wskazane w tej ustawie, i implementujecie przepisy prawa unijnego.

Przyłączając się do tych wszystkich pytań, chciałabym również zapytać, ile w związku z tym szczegółowym nadzorem, znając potrzeby pacjentów, planujecie państwo m.in. na wsparcie dla osób niepełnosprawnych w dofinansowaniu zakupu np. wózków czy innych (Dzwonek) przyrządów ortopedycznych. Dziękuję bardzo, pani poseł. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O udzielenie odpowiedzi na postawione pytania uprzejmie proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana ministra Macieja Miłkowskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! Dziękuję bardzo serdecznie za przedstawione pytania. Tych pytań jest dużo.

W związku z tym nie można stosować reklamy, która jest niewłaściwa.

Pierwsze i ostatnie są trochę niezwiązane, choć związane rzeczowo, to znaczy związane z produktami, wyrobami medycznymi na zlecenie: Jakie będzie dofinansowanie, czy będzie wzrastało dofinansowanie na wyroby medyczne, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? W tym zakresie ta ustawa w ogóle tej sprawy nie dotyczy, ponieważ to jest ujęte w rozporządzeniu w zakresie wyrobów medycznych na zlecenie.

Kiedy będzie finansowane in vitro? To jest nazwa wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, czyli do wszelkich działań laboratoryjnych, produktów.

Tutaj były dyskusje o rejestracji wyrobów medycznych przez firmy, które prowadzą działalność gospodarczą - w związku z tym tam dane osobowe muszą być - jako producent, jako jednostki wprowadzające wyroby medyczne do obrotu. Chodzi o przepisy do sprawowania nadzoru.

One są dookreślone, tak jak państwo wiedzą.

Jak pan prezes urzędu to przedstawił, to jest decyzja administracyjna. Wysokość kary musi być uzasadniona. Od tej wysokości kary można się odwołać. Ale jednocześnie, jak pan prezes bardzo jasno powiedział, w przepisach są ujęte dokładne zasady. Jeśli jest to incydentalne, jeśli jest to naprawione w czasie kontroli - chodzi o te przepisy, które są złamane - wówczas prezes ma możliwość odstąpienia od nałożenia kary w pełnej wysokości. Oczywiście te kary analizowaliśmy.

Trzeba to bardzo mocno uzasadnić.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o wyrobach medycznych zawarty w druku nr 1764 do Komisji Zdrowia celem rozpatrzenia. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii (druk nr 1767)

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić poselski projekt ustawy o powołaniu Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Zgodnie z art. 18 polskiej konstytucji rodzina i małżeństwo, rodzicielstwo i macierzyństwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Wynikające z tego obowiązki państwa mają charakter szczególny, ponieważ zostały zapisane w ustawie zasadniczej, i to w jej pierwszym rozdziale, co wskazuje na ich wagę i pozycję w aksjologii naszej konstytucji.

Dla państwa wynika z nich z jednej strony obowiązek nienaruszania i przeciwdziałania naruszeniom praw rodziny, małżonków i rodziców, a także dzieci wynikającym z działań władzy publicznej, ale także mogących wynikać z działań innych podmiotów, z drugiej strony z tych przepisów konstytucyjnych wynika też konieczność wypełnienia pozytywnego obowiązku w zakresie podejmowania działań służących rozwojowi i dobremu życiu polskich rodzin. To jest konstytucyjna podstawa i zachęta do powołania Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Regulacje naszej ustawy zasadniczej odpowiadają szeroko podzielanemu w Polsce przekonaniu. Zgodnie z badaniami opinii publicznej od lat niezmiennie rodzina należy do najważniejszych wartości dla Polaków. Możemy też powiedzieć, że rodzina i demografia to ostatecznie dwie najważniejsze sprawy dla Polski, nie tylko zresztą dla naszego kraju, ale też dla całej Europy. Jest obecnie oczywiście wiele wyzwań społecznych, gospodarczych i politycznych, w sferze polityki energetycznej, związanych z epidemią koronawirusa, wojną hybrydową na wschodniej granicy Polski, wschodniej granicy Unii Europejskiej, a być może także z głębszymi zagrożeniami geopolitycznymi na wschodzie Europy. Innymi słowy, wyzwań obecnego czasu jest wiele, ale mamy podstawę sądzić, że uda się nam większość z nich przezwyciężyć, w niemałej części w krótkim czasie, a w każdym razie w ciągu kilku lat. Ale wyzwanie demograficzne wydaje się większe, wydaje się mieć zupełnie inną skalę, a ostatecznie ta sprawa, sprawa demografii, wyznacza pozycję i przyszłość społeczeństw i państw, także pozycję i przyszłość Polski i polskiego społeczeństwa. Demografia uzależniona jest od sytuacji i kondycji rodziny. Stąd myśl i potrzeba powołania Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Oczywiste jest, że wzrost demograficzny stanowi podstawowy czynnik zapewnienia trwałości społeczeństw oraz ich rozwoju. Nie ma wątpliwości, że bez tzw. zastępowalności pokoleń w perspektywie kilkudziesięciu lat dochodzi do gwałtownego spadku ogólnej liczby ludności, a tym samym osób czynnych na rynku pracy, co z kolei stanowi chociażby poważne obciążenie dla systemu ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie generuje szereg wyzwań, którym sprostanie wymaga odpowiednich zasobów ekonomicznych i osobowych. Do tego zaś konieczne jest zagwarantowanie wspomnianej zastępowalności pokoleń. W tym kontekście możemy mówić o konieczności podejmowania działań z perspektywą nie na lata, ale na dekady, działań zapewniających bezpieczeństwo demograficzne Polski. Jak dowodzą statystyki i prognozy, bezpieczeństwo demograficzne naszego kraju jest poważnie zagrożone.

W ślad za tym podążą poważne zmiany w strukturze populacji. Programy takie jak 500+ doprowadziły w pewnym stopniu do wyhamowania spadku liczby urodzeń. zwiększyły też poziom bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. ale musimy zrobić więcej. Warto przy tym zaznaczyć, że świadomość konieczności wypracowania spójnej, kompleksowej i długofalowej polityki w zakresie demografii jest komunikowana i podnoszona przez przedstawicieli instytucji rządowych, czego przykładem jest „Strategia demograficzna 2040” Doceniając wagę tego dokumentu, należy - podobnie jak to zrobili jego autorzy - zwrócić uwagę na potrzebę i efektywność działań prodemograficznych prowadzonych w sposób długofalowy i kompleksowy, co potwierdzają doświadczenia takich państw jak Francja, Szwecja czy Węgry. Oznacza to m.in., że osiągnięcie celów demograficznych możliwe jest jedynie wtedy, gdy oprzemy się na rzetelnych i wszechstronnych badaniach naukowych oraz wielowymiarowych działaniach prowadzonych w sposób ciągły i konsekwentny, a więc zapewniający bieżące monitorowanie trendów związanych z szeroko pojętą demografią, a także gdy wypracujemy odpowiednie rekomendacje w celu przeciwdziałania występowaniu negatywnych zjawisk w tym obszarze. Obecnie w Polsce nie istnieje instytucja zajmująca się w kompleksowy sposób badaniem zjawisk demograficznych, zwłaszcza niskiej dzietności, ich wpływu na sytuację społeczeństwa oraz wypracowywaniem adekwatnych sposobów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją.

Francja z problemem, z którym borykamy się dzisiaj w Polsce, borykała się już w okresie międzywojennym, stąd myślenie na ten temat ma tam znacznie dłuższą historię niż w Polsce. Nie ma przy tym wątpliwości, że konieczność konsekwentnego kształtowania skutecznej strategii radzenia sobie z zaistniałym kryzysem jest pilnym zadaniem, od którego realizacji zależeć będzie przyszły poziom życia zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Uważamy, że istnieje konieczność powołania wyspecjalizowanej jednostki zajmującej się kompleksowymi studiami nad procesami zachodzącymi w sferze demografii. Chodzi o instytucję, w której zostanie zagwarantowany odpowiedni stopień niezależności od czynników związanych z prowadzeniem bieżącej działalności politycznej. Jest to niezbędne dla wypracowania właściwych rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki prodemograficznej. Takie instytucje powstały w wielu państwach na świecie: we wspomnianej Francji, ale także w Stanach Zjednoczonych. W naszej części Europy - w Czechach, na Słowacji. na Węgrzech, tak jak pani słusznie powiedziała, pani poseł. Cieszę się, że ma pani taką dużą wiedzę w tym zakresie. Pięknie. Powiedziałem kilka słów o założeniach. które legły u podstaw projektu stworzenia tej instytucji, ale teraz kilka słów o zadaniach instytutu. Zadania instytutu zostały określone w art. 3 projektu ustawy w zakresie umożliwiającym kompleksowe badanie zarówno zjawisk demograficznych, jak i związanych z nimi procesów, oraz wypracowywanie rekomendacji i narzędzi umożliwiających organom państwa prowadzenie odpowiedniej polityki w odniesieniu do pojawiających się wyzwań. Koresponduje to ze „Strategią demograficzną 2040” oraz „Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w której pułapkę demograficzną wskazano jako jedną z najważniejszych barier rozwojowych Polski w najbliższych dekadach. Teraz krótko o tych zadaniach. Po pierwsze, to merytoryczne zaplecze dla trwałej, organicznej polityki prorodzinnej. Po drugie, instytut jest pomyślany jako instytucja naukowa i think tank diagnozujący i prognozujący procesy demograficzne, szanse i zagrożenia, analizujący te procesy wraz z kontekstem kulturowym i ekonomicznym.

Prezes instytutu będzie swoistym rzecznikiem praw rodziny i będzie miał kompetencje analogiczne do innych rzeczników. Będzie uprawniony m.in. do udziału w stosownych postępowaniach wnioskowania o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą oraz inicjowania stosownych zmian w prawie miejscowym.

Nie ma tu żadnych oryginalnych rozwiązań. Wszystkie są tymi.

Jeśli chodzi o ten pierwszy pomysł, to był on wielokrotnie podnoszony przez różne zresztą osoby i środowiska w ramach pracy Rady Rodziny działającej przy minister rodziny.

Ponieważ Polski Instytut Rodziny i Demografii ma łączyć cechy tych dwóch rodzajów instytucji, z jednej strony instytucji badawczej, a z drugiej strony instytucji rzecznikowskiej, ma on posiadać znaczną autonomię. która zapewni niezależność i możliwość prowadzenia swobodnej działalności. Zwrócę też uwagę, że te gwarancje są analogiczne do tych, które posiadają inni rzecznicy: rzecznik praw obywatelskich i rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Ma to być państwowa osoba prawna finansowana z budżetu państwa, z siedzibą w Warszawie, ale z możliwymi oddziałami w kraju, niezależna od organów władzy publicznej zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego, funkcjonująca w sposób ciągły i systematyczny. Prezes instytutu musi być obywatelem Polski, posiadać stopień naukowy, wyróżniać się kwalifikacjami i doświadczeniem z obszaru badań nad rodziną, polityką rodzinną i demograficzną, nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu. W oczywisty sposób nie może być, co wynika z przepisów ustawy, parlamentarzystą.

Kandydat na prezesa instytutu ma być wyłoniony w konkursie przez radę instytutu... ...ani bazar. Konkurs ma mieć dwa etapy: formalny i merytoryczny. Jednocześnie Sejm w określonych przypadkach - w ściśle określonych w ustawie - będzie miał możliwość odwołania prezesa z pełnionej przez niego funkcji. Poza tym wprost w projekcie zagwarantowano prezesowi niezależność od innych organów władzy publicznej tak szczebla rządowego, jak i samorządowego. Instytucją opiniodawczo-doradczą oraz kontrolną będzie rada instytutu, która będzie składać się z dziewięciu członków - pięciu wybranych przez Sejm, dwóch przez Senat, dwóch przez prezydenta.

Już fakt, że Senat wybiera dwóch członków, pokazuje, że tak będzie z pewnością. Ale mam nadzieję, mogę powiedzieć, że ze wszystkich istotnych środowisk politycznych będzie wskazana osoba w radzie instytutu, czyli będą i przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, i przedstawiciele opozycji rekomendowani przez Koalicję Obywatelską, przez ludowców, Lewicę (Dzwonek) czy Konfederację. Jeśli chodzi o jednostki organizacyjne instytutu, które pokazują, czym ma się on zajmować, to: Departament Badań i Analiz, Departament Kultury, Mediów i Edukacji, Departament Współpracy z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi, Departament Współpracy Zagranicznej. Przyjęcie projektowanych rozwiązań spowoduje wydatki z budżetu państwa w kwocie ok. 30 mln zł, natomiast nie spowoduje dodatkowych kosztów finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wysoka Izbo! Jeśli wziąć pod uwagę aksjologię polskiej konstytucji, negatywne trendy demograficzne oraz szereg problemów wynikających z tego rodzaju zjawisk, to powołanie instytutu wydaje się więcej niż wskazane, wydaje się koniecznością niezbędną do wypracowania właściwych rekomendacji i narzędzi w zakresie prowadzenia polityki prodemograficznej. włączając w to prowadzenie długofalowej i systematycznej aktywności nakierowanej na diagnozowanie i kształtowanie trendów społeczno-kulturowych wpływających na kondycję demograficzną Polski. Dziękując za uwagę, proszę o rzeczową dyskusję, w szczególności o unikanie takich argumentów, które w oczywisty sposób są nieprawdziwe, które niejako wynikają z projektu ustawy, które zostały też przeze mnie tutaj przedstawione. Proszę też nie doszukiwać się ukrytych intencji, zamiarów, bo to, myślę, nie służy sprawie. Ostatecznie można powiedzieć, że sprawa demografii jest sprawą ważną dla wszystkich. Tych, którzy mają prawicowe poglądy, lewicowe poglądy, tych, którzy w żaden sposób się nie identyfikują, bo od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja demograficzna Polski. zależy to, jaki będzie los naszego społeczeństwa, po części nas samych, na pewno naszych dzieci. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Dominika Chorosińska. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie złożonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii z druku nr 1767. Z badań socjologicznych jasno wynika, że znaczna część Polaków rodzinę uważa za najwyższą wartość. Synonimem szczęścia indywidualnego jest szczęście rodzinne. Jednocześnie widzimy, że liczba rozwodów z roku na rok wzrasta. Młodzi deklarują, że chcą mieć dzieci, a jednocześnie mierzymy się z ogromnym kryzysem demograficznym.

Ich rola w rozwoju gmin, miast i państw wymaga stałej analizy, badania i opisywania, ponieważ od tej wiedzy zależeć będą kondycja i warunki życia przyszłych pokoleń. Procesy społeczno-kulturowe, demograficzne i ekonomiczne wymagają badania w celu wyjaśnienia i zrozumienia ich współzależności z zachowaniami i dążeniami poszczególnych członków rodziny. Ważne jest, by upowszechniać dobrej jakości wiedzę na temat fundamentalnego znaczenia małżeństwa i rodzicielstwa dla społeczeństwa. The Lancet”, recenzowane, naukowe czasopismo medyczne z Wielkiej Brytanii, jedno z najdłużej wydawanych tego typu czasopism na świecie, twierdzi, że w 2100 r. będzie nas 15 mln. Rodzina od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy była w sercu polityki. To zostało potwierdzone nie tylko słowem, ale i czynem. Aby skutecznie wspierać rodziny, trzeba skutecznie identyfikować problemy, bariery rozwojowe, jeśli chodzi o zakładanie i pomyślne funkcjonowanie rodzin. Takie instytuty działają na całym świecie. Wśród państw Grupy Wyszehradzkiej Polska jest jedynym państwem, które takiego instytutu nie posiada. Klub Prawo i Sprawiedliwość wyraża poparcie dla tej inicjatywy, która wychodzi naprzeciw fundamentalnym wyzwaniom współczesności. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Zgłaszam ten wniosek, ponieważ to nie jest projekt, który ma chronić polskie rodziny i mówić o polskich rodzinach. To jest projekt, który ma tworzyć świat bez różnorodności i bez wolności wyboru. To nie jest projekt ustawy stworzony w trosce o stan demografii w Polsce. To jest projekt, który za 30 mln zł ma promować wybrany przez wnioskodawców konserwatywny, narodowo-katolicki model rodziny i świata.

przez którego kobiety boją się zachodzić w ciążę, bo martwią się o swoje zdrowie, o swoje życie. Instytut rodziny i demografii. Pani Izabela z Pszczyny też miała swoją rodzinę. Trzy najważniejsze elementy tego projektu: superprokurator demograf, edukacja i dane osobowe. Po pierwsze, projekt zakłada, że prezes będzie powoływany na 7 lat i praktycznie będzie nieodwoływalny. Co ciekawe i co jest bardzo trudne do przyjęcia w obywatelskim państwie demokratycznym, superprokurator, prezes instytutu będzie mógł żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych dotyczących rodzin, w sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, będzie mógł brać udział w postępowaniu dotyczącym nawiązania stosunku przysposobienia w sprawach nieletnich. Pytanie brzmi: Po co? Przedstawiciel instytutu będzie mógł dołączyć np. do postępowań rozwodowych. Po to, żeby je utrudniać? Będzie angażował się tam, gdzie akurat ten model rodziny państwu nie odpowiada, bo nie takie małżeństwo, bo rodzina tęczowa, bo nie takie poglądy?

To są realne dzieci, to są realne rodziny. Mamy rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich. Przez lata nie byliście w stanie stworzyć realnej strategii demograficznej w Polsce, przez 6 lat. Rządzicie 6 lat. Instytut ma w tym pomóc? Przez lata nie byliście w stanie zmienić systemu pieczy zastępczej. Nie byliście w stanie stworzyć systemu kontroli przypadków śmiertelnych pobić dzieci w Polsce. Instytut tego nie zmieni. Badania i edukacja. 30 mln zł wykorzystacie nie na badania realne i zgodne z faktami, ale na promocję w szkołach przez organizacje, które będziecie sponsorować z tych pieniędzy, wartości, które odpowiadają wam, które są przeciwne różnorodności, które są przeciwne prawom kobiet, wolności wyboru.

Nie trzeba 30 mln, wiemy, co trzeba robić. Może to państwo w końcu zrobicie. Szanowni Państwo!

Po co? Najintymniejsze szczegóły naszego życia, dane medyczne, edukacyjne, dotyczące stanu cywilnego - po co to w instytucie? No chyba nie po to, żeby wpływać na życie obywateli i mieć intymne informacje o ich życiu. Skoro troszczycie się i powołujecie się na Francję, to: Francja - liberalna aborcja, Francja - edukacja seksualna, Francja - dostęp do antykoncepcji. Może warto pójść tą drogą, a nie tworzyć instytuty. Troszczycie się o rodziny, troszczycie się o dzietność. Mamy na to receptę: żłobki, przedszkola, mieszkania, stabilna praca, partnerstwo w związku. To należy promować.

Pani poseł Wanda Nowicka w imieniu klubu Lewica. Oczywiście, panie pośle. W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy przedstawiam stanowisko dotyczące projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Projekt ustawy jest kolejną inicjatywą posła Wróblewskiego, która przeraża. To za sprawą posła Wróblewskiego Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej uznał, że kobieta musi rodzić, nawet gdy płód ma śmiertelne wady wrodzone i umrze tuż po porodzie. Trybunał Konstytucyjny i osobiście pan poseł Wróblewski ponoszą moralną odpowiedzialność za narażenie Polek w ciąży na utratę życia. O tym zagrożeniu cała Polska przekonała się, gdy umarły panie Izabela z Pszczyny i Anna ze Świdnicy. Ustawa o instytucie rodziny i demografii budzi grozę, bo ma to być jakaś superinstytucja, która ma ogromne kompetencje i pieniądze, a żadnej odpowiedzialności. Otrzymuje uprawnienia innych instytucji, jak Główny Urząd Statystyczny, polityka społeczna, nawet prokuratura. Będzie to instytucja, która wejdzie, powiem kolokwialnie, z buciorami do życia prywatnego Polek i Polaków, by wpływać na nasze życie, zmuszać kobiety do rodzenia interweniować w sprawach rozwodowych albo gdy nastolatki chcą przerwać ciążę. Wtedy w roli prokuratora będzie mógł wystąpić szef instytutu, by zmusić dwunastolatkę do urodzenia wbrew jej woli. Pełna kontrola nad płodnością polskich rodzin. Czy to wciąż science fiction, czy niestety upiorna rzeczywistość, która stanie się faktem, gdy ta ustawa zostanie przyjęta? Przecież nie bez powodu poseł Wróblewski wpisał do ustawy zadanie dla instytutu: uczestnictwo w postępowaniach sądowych w zakresie dotyczącym rodziny lub dzieci na prawach przysługujących prokuratorowi. Przecież instytut posła Wróblewskiego ma zagwarantować więcej urodzin, zatem prokuratorska, czyli oskarżycielska, a nie obrończa, rola w rękach instytutu naprawdę przeraża, bo instytut ma oskarżać. Kogo? Kogo instytut będzie oskarżał? Np. kobiety, które przerwały ciążę w Holandii czy w Czechach, albo lekarza, który przepisał tabletkę „po stosunku”, albo rodziców, którzy zgadzają się na to, by ich córka, zgodnie ze swoją wolą, przerwała ciążę. Ale to nie wszystko. Instytut chce ograniczyć rolę rzecznika praw obywatelskich. Ma być jego kontrolerem i recenzentem. Poseł Wróblewski chce się dobrać za pośrednictwem rzecznika do partii politycznych. Mógłby badać, czy cele i działalność danej partii są zgodne z konstytucją.

Zaangażowanie posłanek Lewicy w inicjatywę obywatelską „Legalna aborcja. Bez kompromisów” pani Przyłębska może uznać za niekonstytucyjne. Dla pani Przyłębskiej nie ma rzeczy niemożliwych. Bez wątpienia prywatność obywateli w praktyce zostanie zniesiona, jeśli ustawa wejdzie w życie, bo instytut mógłby przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań. A jakie dane osobowe są niezbędne do zwiększenia liczby urodzeń? Oczywiście stosowanie antykoncepcji, ciąże i aborcje. I o te dane chodzi panu posłowi, by instytut mógł interweniować i wykorzystywać uprawnienia prokuratorskie przeciwko kobietom i rodzinom. Rozporządzenie o rejestracji ciąż nie wzięło się znikąd. Kontrola nad płodnością kobiet ma być nadrzędnym celem polityki państwa, bo państwo nie tylko chce poznać prokreacyjne decyzje ludzi. Państwo chce w te wybory ingerować. Konstytucyjna ochrona prywatności stanie się fikcją, bo w tym projekcie chodzi o zmuszanie Polek do rodzenia, by realizować demograficzną politykę państwa, by rodziły, choćby miały umrzeć bądź stracić zdrowie. Prezes na otarcie łez i w nagrodę za dręczenie Polek robi z niego nadrzecznika, który będzie mógł wtrącać się w prywatne życie rodzin i będzie mógł urządzać je według swojego widzimisię. A jakie ciągoty ma poseł Wróblewski, to już wiemy. Piekło kobiet to jego dzieło. Jakie będą polskie rodziny? Bez rozwodów, po katolicku, bez praw kobiet.

Pani poseł Bożena Żelazowska w imieniu klubu Koalicja Polska. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawiam stanowisko klubu wobec poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii, druk nr 1767. Tak, panie pośle, rzeczywiście sprawa demografii jest dla nas, Polaków, wszystkich, bardzo ważna. Żyjemy dziś w bardzo trudnym czasie. Zagrożenie kolejnymi atakami hybrydowymi, niedająca się zapomnieć pandemia, rosnące ceny, inflacja. Obiecywaliście tanie państwo. Tymczasem zajmujemy się tworzeniem kolejnej instytucji z siedzibą, zapewne kosztownym zarządem instytutu, radą i pracownikami. Tylko czy od tego wzrośnie dzietność Polaków? Gros jej zadań już dzisiaj realizują samorządy. Czy nie wystarczy naprawdę pomóc tak podobno dobrze funkcjonującemu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej i właśnie samorządom? Rząd rzeczywiście przez 6 lat funkcjonowania nie wypracował długofalowej polityki demograficznej. Nie ma też polityki senioralnej. Nie ma też polityki migracyjnej. Dlaczego cały czas, podkreślam, rząd nie korzysta z doświadczeń samorządów w tym zakresie, chociażby poprzez promocję Karty Dużej Rodziny? Przypomnę, że prekursorem tej karty był burmistrz miasta Grodzisk Mazowiecki kolega Grzegorz Benedykciński. Środki, które możemy przeznaczyć dla polskich rodzin, powinny być dzielone przez gminy, których pracownicy znają sytuację polskich rodzin, powinny być zachętą do rozwoju i posiadania potomstwa. Zawsze jako Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe głosujemy za dobrymi rozwiązaniami dla polskich rodzin. Głosowaliśmy też za programem 500+. Pierwsze programy w tym zakresie zostały wprowadzone, kiedy ministrem pracy i polityki społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. Wtedy powstały takie rozwiązania jak kosiniakowe, wtedy powstały urlopy macierzyńskie, były one wydłużone dla matek. Powstały też liczne, jak państwo pamiętacie, programy dla seniorów. Dzisiaj, drodzy państwo, czas się naprawdę zastanowić, poważnie zastanowić. Czy tworzenie kolejnej kosztownej instytucji zwiększy dzietność Polaków? Czy może potrzebne są inne narzędzia i środki, które sprawią, że w polskich rodzinach będzie rodziło się więcej dzieci? Może warto dofinansować system opieki zdrowotnej, stworzyć mądre rozwiązania dla matek, aby nie bały się zachodzić w ciążę. A przecież jutro będziemy omawiać ustawę o karach dla lekarzy, którzy i tak są w trudnej sytuacji. Często stoją przed wyborem, czy ratować życie, zdrowie matki kobiety.

Brak jest specjalistów w tym zakresie. Dobrze wszyscy wiemy - wielokrotnie był tutaj poruszany ten problem - jak wielki jest brak lekarzy psychiatrów dziecięcych. A tak wiele dzieci cierpi dzisiaj na te schorzenia. Może warto dofinansować pobyt dziecka w żłobku czy przedszkolu. Polskie dzieci, zwłaszcza te wychowujące się w rodzinach mniej zamożnych, na wizytę u specjalisty czekają po kilka albo kilkanaście miesięcy. Potrzebny jest szybki dostęp do stomatologa. Potrzebne są mądre programy wspomagające rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Czy stać nas dzisiaj jako państwo - zadajmy sobie tutaj to pytanie wszyscy - na budowę kolejnej instytucji, która pochłonie. To nie 30 mln, to są kolejne lata funkcjonowania tej instytucji, to będą środki, które będą szły w miliardy. Czy stać nas dzisiaj na to, drodzy państwo? Będziemy się mocno przyglądać waszym działaniom w tym zakresie. Pan poseł Dobromir Sośnierz w imieniu koła Konfederacja. Zapraszam, panie pośle. Pan ma zwolnienie lekarskie. 30 mln zostanie zabrane pracującym rodzinom i przekazane na instytut zadumy nad demografią. Co w tym pomyśle może pójść nie tak? To szaleństwo powoływania kolejnych instytutów ma być według rządu PiS, jak rozumiem, odpowiedzią już na każdy kolejny temat. Pan Wróblewski mówił o Czechach i Francji. Jeśli są tam takie instytuty, to może po prostu taniej będzie odkupić od nich te rozwiązania? Tak że może sporo zaoszczędzimy. Jeśli potrzebujecie jakiejś ekspertyzy, to można ją zamówić na rynku za, nie wiem, 50 tys., powiedzmy, a nie 30 mln. Biurka i etaty to nie jest odpowiedź na problemy demograficzne. Albo ja wam pomogę za 1% tej sumy. Dzisiaj nawet za darmo wam powiem o tym, co jest nie tak z demografią. Oczywiście na część z nich nie mamy i nie będziemy raczej mieli większego wpływu, np. upowszechnienie się antykoncepcji, wbrew przekonaniu pani posłanki Rosy, albo emancypacja kobiet. To są zjawiska, które z całą pewnością osłabiają przyrost demograficzny w każdym kraju, w którym występują, ale raczej nic na to się nie poradzi. Systemy emerytalne przede wszystkim. Jednym z powodów, dla których ludzie posiadają dzieci i zawsze posiadali dzieci, było zabezpieczenie na starość. Zniedołężniali starcy byli utrzymywani przez dzieci i wnuki. Przekonanie o konieczności posiadania dzieci zostało zapisane w dawnej kulturze, która wysoko ceniła sobie rodzicielstwo, płodność, więzi rodzinne. Analogicznie przerwanie przez pobismarckowskie reżimy socjalne związku między posiadaniem dzieci a utrzymaniem na starość doprowadziło do przemian kulturowych zmierzających w przeciwnym kierunku, czyli do rozpadu więzi rodzinnych, do coraz wyraźniejszego postrzegania dzieci jako raczej problemu, a nie daru Boga. Rozwiązanie: likwidacja przymusu ubezpieczeń emerytalnych. Państwowa edukacja. Państwo rzuca na rynek edukację, którą nazywa darmową, ona de facto jest przedpłacona w podatkach. Wszystko, co darmowe, jest nadużywane, więc uruchomiono w ten sposób absurdalny wyścig zbrojeń, w którym edukację rozciąga się już niemal do trzydziestki, pomimo że większość ludzi zupełnie jej nie potrzebuje, bo wykonuje proste prace, do których mogliby się przygotować w tydzień czy w miesiąc. Każdy chce mieć jak najwyższe wykształcenie - skoro to nic nie kosztuje - żeby się lewarować na rynku pracy, ale ponieważ robią to wszyscy, te wysiłki i tak się równoważą. To również powoduje przemiany kulturowe: powstanie nowego etosu przedłużonej niedojrzałości, hedonizmu młodzieńczego i w rezultacie odsuwanie ojcostwa i macierzyństwa w czasie. Rozwiązanie: gruntowa deregulacja i prywatyzacja edukacji. Podatki - trzecia sprawa. Wysoki klin podatkowy i sztywna regulacja rynku pracy dotykają najbardziej młodych ludzi. Zabiera się im pieniądze, kiedy są młodzi, zniechęcając do posiadania dzieci, żeby oddać w późniejszym czasie w postaci różnych programów socjalnych i emerytur. Upaństwowienie małżeństw, ułatwienie rozwodów i ingerencja w wychowywanie dzieci odbierają rodzinom, ludziom poczucie sprawczości. Coraz bardziej ludzie czują, że wychowują podatników dla chciwego państwa, a nie własne dzieci zgodnie z własnymi poglądami. Wspieranie samotnych matek powoduje, że jest więcej samotnych matek i rozbitych rodzin. To wszystko również zapisuje się w kulturze i przebudowuje nasze wyobrażenia o tym, jak powinno wyglądać nasze życie. Rozwiązanie: odczepienie się państwa od rodziny, przywrócenie pełnej wolności w wychowywaniu dzieci. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Na tej sali oglądaliśmy już wiele szkodliwych projektów, jednak ten jest wyjątkowy w specjalny sposób. Bo to nie jest druk, to jest weksel, który skrajnie radykalna frakcja Zjednoczonej Prawicy wypisała na 30 mln rocznie i położyła przed Jarosławem Kaczyńskim. Płać za ich wierność negocjowalnego afektu, bo inni dostali, a oni - jeszcze nie. Bo kiedy prezes miał ochotę iść z opozycją bardziej na ostro, wnieśli haniebny wniosek do tzw. Trybunału Konstytucyjnego, który skończył się piekłem dla polskich kobiet i śmiercią Izabeli z Pszczyny. A teraz my, podatnicy, zapłacimy za ich chore urojenia, które wyglądają tak, jakby pisali je nie polscy posłowie, ale sponsorowani przez Kreml fundamentaliści. Pod nazwą Polski Instytut Rodziny i Demografii nie kryje się nowa instytucja dbająca o podstawową komórkę społeczną, a trybunał inkwizycyjny, który będzie miał uprawnienia prokuratorskie. W połączeniu z rejestrem ciąż to będzie prawdziwy młot na prawa kobiet, na wolności obywatelskie i faktyczne dobro rodziny. I to narzędzie dajecie do ręki ludziom, którzy otwarcie kwestionują nasze prawa. Ten instytut to de facto instytucjonalizacja skrajnego radykalizmu w Polsce i wciągnięcie marginalnych środowisk do rządzenia. Pamiętajcie o jednym: te środowiska koniec końców i was skonsumują. Sami staniecie przed ich trybunałami. 30 mln zł na początek to cena, za jaką sprzedajecie bezpieczeństwo kobiet w Polsce. Tworzycie brutalną policję obyczajową do walki z kobietami - z armią pseudoprokuratorów, którzy będą ścigać za, tu cytat, naruszenie praw lub dobra dziecka. Przypomnijmy, że dla posła Wróblewskiego, głównego inicjatora tego arcydzieła, definicję tę spełnia ciąża z kazirodztwa lub gwałtu, ale również taka, która zagraża życiu matki. A więc o ile lekarze po wyroku TK boją się pomagać kobietom, o tyle teraz będą mieli w pamięci realną groźbę cywilnego procesu, jaki będzie mógł im wytoczyć ten IPN do spraw dzieci za ratowanie życia przyszłej matki, kiedy ciąża obumiera. Jako Polska 2050 składamy wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Stanowczo sprzeciwiamy się szarganiu takich pojęć jak „nauka” i „dobro publiczne” dla chwilowego zaspokojenia apetytów radykałów na kasę, władzę i możliwość zastraszania polskich kobiet. Wasz instytutu demografii i rodziny to będzie groteska dla całej Europy.

Bo tak właśnie będzie to wyglądało: jak kabaret transmitowany na cały świat, gdy radykałowie pokroju Bartłomieja Wróblewskiego, Kai Godek i eksperci Ordo Iuris będą oceniali polskie rodziny. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Szramka w imieniu koła Polskie Sprawy. Wysoka Izbo! Mam wrażenie, że niektórzy na siłę próbują na nowo odkryć Amerykę. Nie pamiętam, żeby w którejkolwiek z tych ankiet w kwestii dzietności, kwestii rodziny na pierwszym miejscu pojawiało się to, że największą potrzebą Polaków jest stworzenie instytutu rodziny i demografii. Szanowni Państwo! Wystarczy wsłuchiwać się w ten głos Polaków i odpowiadać na te potrzeby. Zapewniam was, że instytut to nie jest najważniejsza potrzeba Polaków. Polskie rodziny potrzebują niskich podatków, potrzebują przejrzystego, prostego, przyjaznego prawa, a przede wszystkim potrzebują tego, żeby politycy aż z taką nachalnością nie wchodzili z butami w ich życie. Jeśli macie przekonanie, że ten instytut cokolwiek naprawi, to dlaczego nie pójdziecie dalej i nie stworzycie instytutu szczęścia, zdrowia i dobrobytu po to, żeby sprawił, że wszyscy będziemy zdrowi, szczęśliwi i będziemy mieli dobrobyt? Faktycznie, może lepiej tego nie podsuwać. Uznajmy, że tego nie mówiłem. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas - 1 minuta. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Trzeba powiedzieć, że to dobrze, że w końcu rozmawiamy o sprawie tak istotnej jak demografia, zastępowalność pokoleń, i to nie tylko okazjonalnie, ale w aspekcie powołania nowej instytucji - Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Tego, jak jest to ważne w aspekcie rodziny, rozwoju społecznego i gospodarczego i przyszłości Polski, dowodzą statystyki i prognozy, z których wynika, że bezpieczeństwo demograficzne Polski jest poważnie zagrożone. Dlatego dobrze, że w sposób systemowy, przez Polski Instytut Rodziny i Demografii będziemy mogli najpierw badać procesy zachodzące w rodzinach i w społeczeństwie, a następnie szukać rozwiązań najlepszych dla rodziny. Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni Politycy PiS! Mówiliście kiedyś: może kradniemy, ale się dzielimy, a teraz przestaliście się nawet dzielić. Bo jaki zysk ma mieć polska rodzina z tego, że będziecie dublować zadania rzecznika praw dziecka, licznych instytutów zajmujących się dzietnością i demografią oraz ministerstwa polityki społecznej? Jaki to ma sens, oprócz przytulenia pieniędzy dla swoich? Chyba jeden. Otóż obsesjonaci będą mogli grzebać w łóżkach polskich rodzin, będą mogli kontrolować, czy rodzice wychowują swoje dzieci zgodnie z waszymi wartościami, a nie z wartościami zgodnymi z konstytucją. Wielka prośba od większości polskich rodzin: przestańcie im szkodzić. Pan Wróblewski powiedział, że polska rodzina potrzebuje instytutu. Bzdura na resorach.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! To kolejny projekt ustawy w sprawie powołania nowej instytucji publicznej, bardzo kosztownej. 30 mln, ale o tym później. W art. 10 w ust. 1 czytamy, że kadencja prezesa instytutu wygasa w razie śmierci, rezygnacji, odwołania, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wnioskodawcy! Oprócz podstawowego pytania, dla kogo te nowe posady, mam pytanie: Czy stanowisko prezesa ma być dożywotnie? Może te 30 mln warto przekazać na leczenie niepłodności.

To jest np. 7 tys. zabiegów in vitro. Pan poseł Krystian Kamiński, Konfederacja.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przez te 5 minut zdążyłem trochę zweryfikować ten temat. W związku z tym mam pewne wątpliwości, czy taki instytut jest rozwiązaniem w zakresie dzietności gdziekolwiek, tym bardziej że jeśli brać pod uwagę rdzenną ludność Francji i tę napływową, to już w ogóle ta dzietność poszła w dół całkowicie. Miałbym wiele pytań odnośnie do tego instytutu, bo całkowicie nie przekonuje mnie to, co państwo mówili, ale jeśli słyszę, że problemem demografii jest aborcja i antykoncepcja, to po prostu trzeba jedno stwierdzić: ta cała lewicowo-liberalna opozycja to jednak stan umysłu. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy patrzę na proponowane uprawnienia prokuratorskie nowego prezesa, to chyba wiem, o co chodzi państwu posłom wnioskodawcom. Chcecie wystraszyć ludzi już tak na amen. Chcecie powołać nowego urzędnika, który będzie takim naturalnym środkiem antykoncepcyjnym. Jak ludzie sobie pomyślą, że będziecie ich ścigać, ciągać po sądach, to na pewno dwa razy zastanowią się na tym, czy chcą mieć potomstwo. Tu jest też drugie dno. Jeżeli rząd PiS z czymś sobie nie radzi, tak jak z demografią, to powołuje za publiczne pieniądze taki instytut z kadrami pełnymi zaufanych działaczy i rodzin Prawa i Sprawiedliwości i prowadzi działalność propagandową, która tę nieudolność rządu ma przykryć. To właśnie będzie robił ten instytut. Ustawa jest do odrzucenia, to oczywiste. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Koleżanki i Koledzy z partii rządzącej! Rządzicie już ponad 6 lat, wprowadziliście bardzo wiele programów, w ramach których na sztandarach mieliście rodzinę, demografię, dobro polskich rodzin, a jakoś demografia nie skoczyła do góry. Jesteśmy na tym samym poziomie, na jakim byliśmy, kiedy wchodziliście do rządu. Pytanie: Czy wy zadajecie sobie pytanie, co robicie nie tak? Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Bezapelacyjnie dzisiaj żyjemy w czasach największego ataku środowisk lewackich na rodzinę. od czasów rewolucji październikowej w Rosji w 1917 r., kiedy to komuniści sowieccy próbowali rozwiązywać rodziny i wprowadzać nowe modele współżycia społecznego. Bardzo dziękuję za projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii, niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w 2012 r. ówczesny Klub Parlamentarny Solidarna Polska wystąpił z projektem ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny. Ta ustawa została odrzucona w pierwszym czytaniu głosami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Ruchu Palikota. Tylko Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska była za, bo my jesteśmy za rodziną, bo my jesteśmy za prawami rodziny.

Deklarowanym powodem powstania tej ustawy jest zbadanie tego, jak doszło do tej zapaści demograficznej w Polsce. Gdybyście użyli aparatu umysłowego, to bardzo szybko byście się zorientowali, że to wasza przemyślana polityka doprowadziła do zapaści demograficznej w Polsce. Po pierwsze, jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, których absolutnie zainspirował saudyjski urząd komitetu krzewienia cnót. A drugi realny powód jest taki, że pozazdrościliście prezesom i zarządowi Polskiej Fundacji Narodowej i innych tego typu organizacji i chcieliście mieć do wydania 30 mln.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Dzisiaj Sejm powołuje policję obyczajową do walki z Polkami na czele z superprokuratorem. Instytut będzie miał zagwarantowany pełen wgląd w nasze dane, nawet te wrażliwe, zatem medyczne i intymne. Rejestr ciąż Polek będzie monitorowany przez ten instytut. A ja mam do was pytanie: Czy każdy Polak będzie miał swoją teczkę w tym instytucie? Jak wy nie wiecie, na co wydać 30 mln zł, to Polacy wam mówią: wydajcie je na żłobki, przedszkola, wydajcie je na in vitro. Ale wam powiem dalej: dzisiaj poseł sprawozdawca z tego miejsca powiedział, że szefem tego instytutu nie będzie mógł być rozwodnik. Otóż kwestią dotyczącą rodziny zajmujcie się na swoich zebraniach partyjnych, a nie nudźcie Polaków tym tematem. Polacy sami wiedzą, jak ma wyglądać ich rodzina.

Pan poseł Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie Pośle Wróblewski! Przedstawiony przez pana projekt ustawy przewiduje bardzo szerokie kompetencje prezesa instytutu. Media donoszą, że to pan zostanie nagrodzony tym stanowiskiem. Pierwsze pytanie: Czy to jest prawda? Słynie pan z fundamentalistycznych religijnych poglądów, popierał pan wręcz z radością bestialski wniosek, którego akceptacja przez pseudo-TK doprowadziła do śmierci. Szanowni państwo, czy naprawdę wyobrażacie sobie, aby poprzeć projekt, który pozwoli prezesowi instytutu uczestniczyć we wszystkich postępowaniach sądowych, w których biorą udział obywatele? Jakie poglądy będzie prezentował podczas tych postępowań? Czy podczas rozpraw będzie mówił np. ofiarom przemocy, że obowiązkiem kobiety jest dbanie o męża? Czy bitemu dziecku powie, że tylko pełna rodzina zapewni mu rozwój? Czy ofierze pedofilii powie, że sama lgnęła do sprawcy albo że to jest bioenergoterapia?

W art. 11 tej niebezpiecznej dla kobiet, małżeństw, par ustawy prezes instytutu rodziny i demografii uzyskuje uprawnienia prokuratorskie na skalę większą niż np. prezes NIK. Może zasięgać informacji, w tym wrażliwych danych osobowych, z każdej organizacji, instytucji, organu administracji publicznej. Nie sądzę, że prezes - bo zanosi się na to, kim będzie prezes, a na pewno na to, jakie cele będzie realizował - nie będzie też ewidencjonował nie tylko ciąż, ale i środków antykoncepcyjnych. Czy według projektodawców będzie tam baza danych, kto, jaka para.

Wysoka Izbo! To, że Lewica jest przeciwko, to nie dziwi, nie jest to nic nadzwyczajnego. Debata jak debata, powiedziałbym, normalna w Izbie. Ale mam pytanie do posłów z Konfederacji. Czy jesteście za demografią, czy jesteście przeciwko demografii? Czy może czas najwyższy powiedzieć wprost i szczerze, że wam się to nie podoba, dlatego że jest to nie wasza ustawa, i czas nie grać, tylko powiedzieć, czy jesteście za rodziną, czy jesteście za demografią? Pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Panie pośle Szłapka, pan już był na mównicy, wykrzyczał się, wygroził, więc może teraz spokojniej posłuchać proszę. Normalna. Nie, jeśli krzyczy z ławy sejmowej, zachowuje się w ten sposób, to nie jest właściwe zachowanie i zwracam uwagę. Bardzo proszę, pani poseł. PiS powołuje instytut rodziny i demografii, który ma zachęcić Polki do rodzenia dzieci. Ma kosztować 30 mln rocznie, będzie miał prezesa z prokuratorskimi uprawnieniami i 7-letnią kadencją, którego trudno też będzie odwołać. Prezes będzie miał też do pomocy dziewięciu członków rady, a wszyscy oni będą sowicie wynagradzani. Chcecie zatrzymać depopulację? Chcecie zażegnać zapaść demograficzną w Polsce? Chcecie, by Polki rodziły więcej dzieci? To dajcie nam, Polkom, żyć w spokoju, nie wchodźcie z buciorami do naszych sypialni, nie zaglądajcie do naszego życia i nie zabierajcie nam prawa do decydowania o sobie. Mam pytanie do przedstawiciela wnioskodawców Bartłomieja Wróblewskiego, który zgotował Polkom piekło kobiet, zdaje się, też przyszłego prezesa tego instytutu. W jaki sposób instytut ma egzekwować założenia rządowej Strategii Demograficznej 2040, której, po pierwsze, jeszcze nie ma, a która, po drugie, jest ostro krytykowana przez środowiska naukowe, przez socjologów, demografów, ekonomistów (Dzwonek), za skrajną ogólnikowość merytoryczną i przeładowanie ultrakonserwatywną ideologią? Ponad jakimi podziałami powstał ten projekt? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Droga prawa strono sceny sejmowej, tak dużo i tak pięknie mówicie o rodzinie, że aż mam ochotę zapytać, ilu jest po waszej stronie rozwodników i ile macie dzieci. Używacie wielkich, okrągłych słów o świętości polskiej rodziny. Chcecie dać uprawnienia prokuratora rodziny właśnie po to, żeby zaglądał w miejsca intymne, żeby zaglądał kobietom pod kołdrę. Wasza polityka społeczna, wasza polityka prorodzinna jest tak bardzo nieskuteczna, że musicie dzisiaj doić państwo na 30 baniek dodatkowym instytutem. Bo gdyby była skuteczna, ten instytut byłby niepotrzebny. Panie pośle Wróblewski, w 2017 r. napisałam do pana wiadomość, kiedy złożył pan wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a pan odpowiedział i złożył pan pewną deklarację: Byłem jednym z wnioskodawców programu „Za życiem”, który wspiera matki i rodziny dzieci niepełnosprawnych. Takie działania będę kontynuował w przyszłości. To jedna z tych rzeczy, z których pan się nie wywiązał, i to jeden z tych argumentów, dzięki którym wiemy dzisiaj na pewno, że ten instytut także na pewno się nie uda. Zapraszam. Wysoka Izbo! Ja osobiście bardzo się cieszę, że powstanie taka instytucja jak instytut rodziny i demografii. która w sposób profesjonalny, naukowy, fachowy będzie wspierać polskie państwo w oddziaływaniu na procesy demograficzne i będzie wspierać polskie rodziny. W projekcie ustawy projektodawcy nakreślili bardzo wiele celów instytutu. Chodzi o przygotowywanie analiz, ekspertyz, studiów prognostycznych, zgłaszanie propozycji rozwiązywania problemów. Jednocześnie w uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje się, że jeśli nic się nie zmieni, to do roku 2050 liczba ludności naszego kraju zmniejszy się o 4,5 mln. Moje pytanie w związku z tym jest takie: Czy powstanie instytutu może przyczynić się do zmiany tych bardzo niekorzystnych trendów? Dziękuję. Pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Zawsze wiedziałam, że PiS-owi marzy się wielka inkwizycja z wielkim inkwizytorem - panem Wróblewskim. Nie mam żadnych wątpliwości, że to coś między prokuraturą a policją moralną i ma służyć jednemu - żeby zaglądać Polakom do łóżka i patrzeć, jak żyją.

Pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Kaczyński! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ludzie decydują się na potomstwo, gdy czują się bezpiecznie. Kiedy w ich kraju jest stabilna sytuacja ekonomiczna i nie ma szalejącej inflacji. Gdy opieka medyczna chroni zdrowie i życie kobiety. Gdy inwestuje się w najnowsze metody leczenia niepłodności, w tym in vitro. Gdy każde dziecko, nawet w najmniejszej wsi, od urodzenia ma dostęp do żłobka, a potem do przedszkola. Gdy kobiety mają równe szanse na rynku pracy. Gdy rodzice mogą wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi wartościami, nie waszymi. Gdy państwo dba o środowisko, o czyste powietrze, wodę, inwestuje w zieloną energię, nie wycina lasów i troszczy się o zdrowie przyszłych pokoleń. Gdy rząd prowadzi pokojową politykę, dba o sojusze i dobre stosunki. A wy robicie wszystko odwrotnie (Dzwonek), dlatego kraj się wyludnia. Chcecie, żeby Polki rodziły? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przykro się słucha tych słów. padających ze strony opozycji, polskich posłów.

Dziwią mnie te głosy sprzeciwu - sama nie wiem przeciwko czemu. Przeciwko rodzinie? Czy przeciwko dzieciom? I ta mizerna próba zrobienia na czymś bardzo dobrym, co już dawno powinno zaistnieć w Polsce, polityki i ta chęć chwilowego zaistnienia w mediach. Opozycja mówi o aborcji - po to przyszliście do Sejmu, żeby podejmować działania umożliwiające zabijanie przyszłych pokoleń? Każde życie powinno być otoczone opieką i szacunkiem, podobnie jak rodzina. Te działania od samego początku podejmuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast fałszywość działań opozycji (Dzwonek) jest ewidentna. Z jednej strony mówi o demokracji i równouprawnieniu, dbaniu o kobiety, o konstytucyjne prawa naszego społeczeństwa.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Polski Instytut Rodziny i Demografii brzmi dumnie, prawda? Oto polski rząd dba o polskie rodziny i chce chronić społeczeństwo przed niżem demograficznym. Wszyscy wiedzieliśmy, że to nie zadziała i nie zadziałało, a rząd teraz mówi: nie, nie taki był cel tego programu. W imieniu rodzin chcecie całkowicie zakazać aborcji. Czy ma to wpływ na demografię? Tak, ma, bo kobiety boją się po prostu zachodzić w ciążę. Niestety nie dla was, bo przecież najważniejsza jest ideologia. Ten instytut to jedynie fasada, na której chcecie budować swoje rzekome przywiązanie do tradycji i do wartości. Dziękuję. Pani poseł Agata Katarzyna Wojtyszek, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku wspierał i wspiera polskie rodziny. Jest wiele programów, na które według was nie było pieniędzy, tak jak na program 500+. To ten program wyciągnął ze skrajnej biedy polskie dzieci i polskie rodziny. Pozytywny wpływ wychowania w rodzinie jest związany przede wszystkim z realizowanymi w rodzinie wartościami, wzajemną więzią uczuciową, pełnionymi w rodzinie rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. Dobrej rodziny w procesie wychowania i wzrastania dzieci i młodzieży nie jest w stanie zastąpić nikt, dlatego polityka państwa, polityka instytucji samorządowych, instytucji pozarządowych powinny być nakierowane na pomoc udzielaną rodzinie i w rodzinie. Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania (Dzwonek) i rozwoju dziecka.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Instytut ma być zapleczem polityki prorodzinnej i prodemograficznej. Mam zatem pytanie: Jakie rozwiązania będzie wprowadzał instytut, skoro flagowy program „500+” nie przyniósł wzrostu liczby urodzeń? Czy to mają być takie rozwiązania, jakie proponujecie dotychczas, czyli nakazy, zakazy i kary? Pseudowyrok TK skazujący kobiety na cierpienie i śmierć. Wprowadzenie cnót niewieścich, najlepiej przed trzydziestką, aby rodzić dzieci, a nie zajmować się rejestru ciąż, całkowity zakaz aborcji pod karą 25 lat więzienia, wprowadzenie utrudnień przy rozwodach. Planujecie nawet zmniejszenie liczby cięć cesarskich przy porodach. I na koniec prezes instytutu, który będzie miał uprawnienia prokuratorskie. Po co? Po to, by ścigać i karać kobiety. Fanatyzm zabija. Nie trzeba powoływać instytutu i wydawać 30 mln na to, aby stwierdzić, że kobiety boją się i dalej (Dzwonek) będą się bać zachodzić w ciążę. Wkrótce w Polsce zachodzić będzie, ale już tylko słońce. Pan poseł Kazimierz Moskal, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Każda ustawa na pewno wywołuje różnego rodzaju emocje. Każdą ustawę można skrytykować. Z tym że moje oczekiwanie zawsze było takie, żeby, jeżeli jest projekt ustawy, odnosić się do pewnych rozwiązań, które są w tej ustawie. Natomiast zadajmy sobie pytanie, na ile wyrażamy swoje poglądy polityczne czy etyczne, a na ile odnosimy się do tej ustawy.

Mam też takie pytanie: Czy prezes instytutu, czy rada instytutu jest zabarowana dla ludzi prawicy, czy też każdy może startować w tych wyborach i konkursach?

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Najpierw wypadałoby zadać pytanie, gdzie jest minister do spraw rodziny. Skoro jej nie ma, być może rząd nie popiera tego projektu. Cieszę się, że jest pani pełnomocniczka rządu do spraw polityki demograficznej, niedawno dowiedziałem się, że od 2 lat jest takie stanowisko w rządzie. Jest również Rada Rodziny - nie wiem, czy państwo wiecie - w skład której wchodzi troje posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze mało? Potrzebny jest instytut. Szanowni państwo, to będzie 36. instytut, agencja rządowa, czy też fundusz. Od 30 mln zł na Fundusz Patriotyczny nie przybyło w Polsce patriotyzmu. Przybyło więcej nienawiści, więcej dzielenia i ksenofobii. Od tego instytutu również nie przybędzie lepszej polityki demograficznej. Chodzi tak naprawdę o to, żeby zagospodarować te 30 mln.

Wznawiam obrady. Pytanie zadaje pani poseł Beata Strzałka, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Na liczebność i strukturę ludności wpływają płodność, umieralność, migracja i zmiany kulturowe. Współczesny model rodziny, zmiany priorytetów, odraczanie decyzji o posiadaniu dziecka znacząco wpływają na demografię również w Polsce.

Jako społeczeństwo mamy coraz większą świadomość, że należy wypracować kompleksowe rozwiązania, badania i politykę w zakresie demografii. Konieczne jest zagwarantowanie warunków do tworzenia i funkcjonowania rodzin, które urodzą i wychowają kolejne pokolenia. W związku z tym chcę zapytać, jakie zadania będą realizowane przez instytut w tym obszarze. Pani poseł Jagna Marczułajtis-Walczak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Polityka demograficzna to jest największa klęska rządów PiS. Nie pomogło 500+ i nie pomoże kapitał opiekuńczy. Od 6 lat systematycznie i konsekwentnie niszczycie polską demografię i poczucie bezpieczeństwa polskich kobiet. Zlikwidowaliście in vitro, zaostrzyliście prawo do przerywania ciąży, planujecie utrudnić i wydłużyć procesy rozwodowe. Efekty waszych działań są tragiczne. Pani Izabela z Pszczyny nie żyje, a wiele młodych ludzi boi się zakładać rodziny i rodzić dzieci. Ten instytut to kolejny program stołek+ w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast (Dzwonek) tworzyć kolejną instytucję, lepiej stworzyć program wsparcia kobiet i rodzin oparty na poczuciu wolności, poprawie standardów okołoporodowych, zwiększeniu bezpieczeństwa i opieki nad ciężarnymi w Polsce i na to przeznaczyć środki finansowe. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! poprą, panie pośle, tak, kluby opozycyjne. Dlaczego? Demografia to jest najważniejsza sprawa w rozwoju Polski, również gospodarczym. Przedmówczyni powiedziała tutaj o 30 mln zł i w każdym przemówieniu to się powtarzało: 30 mln zł. A więc mam pytanie: Czy to za waszych rządów wydano 50 mln zł na portal internetowy dla bezdomnych, tak by każdy z nich miał laptopa lub telefon komórkowy? Pomyślcie najpierw o tym, jak wyście wydawali pieniądze. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo! Demografia w Polsce woła o pomstę do nieba. W ciągu ostatniego roku urodziło się 334 tys. dzieci, a zmarło 538 tys. Polek i Polaków.

To jest fiasko waszej polityki. Potrzebna jest prawdziwa polityka, a nie tworzenie pseudoinstytutu jak w komunie.

Dodatkowo jeszcze chcę powiedzieć, że ten projekt jest niekonstytucyjny, gdyż zmusza rzecznika praw obywatelskich do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Takie uprawnienia ma szef tego instytutu. Pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Jest pan poseł? Pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiecie państwo, dlaczego spada poczucie bezpieczeństwa kobiet, które miałyby rodzić dzieci w Polsce? Bo coraz bardziej chcecie ingerować w nasze życie. Chcecie wchodzić z butami do naszych domów, zaglądać do łóżek, mówić, co mamy myśleć i co mamy robić. Powołacie kolejny instytut za 30 mln zł z niemal nieodwoływalnym prezesem, który będzie miał uprawnienia prokuratorskie. 30 mln zł na analizy dotyczące dzietności Polaków. W tym pewnie znowu będą gigantyczne wynagrodzenia dla prezesa, prawda, panie wnioskodawco? Wiecie co można zrobić za te pieniądze? Można realnie działać. Wy moglibyście zrealizować trzy takie programy w ramach tego budżetu i to byłoby realne wsparcie rodzin i wsparcie rozwoju dzietności w Polsce. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Bartłomiej Dorywalski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Tyle razy usłyszeliśmy na tej sali wypowiedzi na temat instytucji trybunału inkwizycyjnego, inkwizycji. Ale jak jest inkwizycja, to i heretycy muszą być. Szanowni państwo, przecież te zapisy, gdy sprawdzamy Kodeks postępowania administracyjnego, znany przecież państwu, są w naszym prawie od ponad 60 lat, jeśli chodzi o udział prokuratora. Zachęcam do lektury. Art. 143 i 144 k.p.a., wersja z roku 1960. Przecież te przepisy obowiązują do dziś. Art. 183 Kodeksu postępowania administracyjnego. Prokurator ma prawo, nie obowiązek, żądać wszczęcia postępowania i wziąć udział w toczącym się postępowaniu. Ale w jakim celu? W celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. Jeżeli państwo tak uderzają w ten przepis, to czy państwo stoją na granicy prawa, na straży prawa czy na straży (Dzwonek) bezprawia? Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pierwsza moja pacjentka sprzed 45 laty na oddziale szpitalnym to kobieta, która miała czworo dzieci, a 14 zabiła, 14 aborcji wykonała. Dostrzegam fałszywą troskę ze strony kobiet tutaj, na sali, i matek z opozycji, ponieważ widzę, że domagacie się poszerzenia wskazań do aborcji pewnie na życzenie. Czy państwo wiecie, co jest główną przyczyną wrogości ludzi wobec dzieci i siebie? Brak szacunku do życia ludzkiego. Instytut chce pomagać rodzinie. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Słyszę od lewicowych posłanek, że instytut rodziny i demografii zabierze Polkom i Polakom rozwody. Tymczasem rozwód dla większości małoletnich dzieci rozwodzących się rodziców to nie jest żadne dobrodziejstwo, tylko największa życiowa tragedia. Dlaczego moi rodzice się rozwodzą? Takie pytanie zadaje sobie wiele dzieci, których rodzice postanowili zakończyć związek małżeński. Rozwody mają olbrzymie skutki ujemne nie tylko dla dzieci, ale także dla społeczeństwa, a nawet dla gospodarki państwa. Nie, instytut rodziny i demografii nie zlikwiduje rozwodów i takich pomysłów nie ma.

Instytut nie zlikwiduje też aborcji, antykoncepcji, nie będzie (Dzwonek) zaglądał do łóżka, nie będzie zabraniał kobietom robić kariery, ale będzie działał tak, aby te Polki, które chcą robić karierę, a jednocześnie chcą mieć dzieci, mogły te dwie rzeczy połączyć z korzyścią dla siebie, dla dzieci i dla swojej rodziny. Do wnioskodawcy mam pytanie: Czy instytut rodziny i demografii będzie miał inicjatywę ustawodawczą, tak jak boją się tego posłanki Lewicy? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej panią minister Barbarę Sochę. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Chciałam powiedzieć kilka zdań na temat tego, o czym była dzisiaj mowa na tej sali, czyli kwestii związanych z demografią i projektem poselskim dotyczącym powołania Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Przysłuchiwanie się tej debacie jest jednym z argumentów za tym, że potrzeba nam szerokiej edukacji i wiedzy na temat zjawisk demograficznych. Ministerstwo, panie pośle, ma swoje zadania, które panu jako posłowi są doskonale znane i nie trzeba ich tłumaczyć.

Jeśli chodzi o kwestie związane z edukacją i znajomością procesów demograficznych, to uważam, że my wszyscy tutaj jako osoby, które mają wpływ na stanowienie prawa, na legislację w tym kraju, jesteśmy zobowiązani do tego, by mieć podstawową wiedzę w tym zakresie.

Absolutnie nie jest prawdą to, co dzisiaj padało kilkakrotnie - że w ubiegłym roku urodziło się w Polsce najmniej dzieci. To jest nieprawda. To są osoby, które w tym roku poszły na studia. To jest nasze najnowsze młode pokolenie, które już zaczyna wchodzić na rynek pracy, wejdzie na niego w 100% za 5 lat, i to są najmniej liczne roczniki w historii powojennej Polski. Co to oznacza? To oznacza dwie rzeczy, szanowni państwo. Po pierwsze, urodziło się wtedy najmniej dzieci, mimo że było relatywnie dużo kobiet, które mogły rodzić, było ich ponad 10 mln.

To jest największa tragedia i katastrofa demograficzna.

Demografowie od 20 lat apelują o stworzenie odpowiednich instytucji, które skoordynują polityki w tym zakresie. Przekonanie, że jeden instrument, nawet taki radykalny, kosztowny i duży, jakim jest program 500+, miałby odwrócić trendy demograficzne, najlepiej świadczy o braku elementarnej wiedzy w zakresie demografii. Francuski instytut studiów demograficznych INET to instytucja, która od 70 lat prowadzi analizy, projektuje polityki, gwarantuje ciągłość wiedzy każdemu kolejnemu rządowi francuskiemu.

Przecież nie będziemy rządzić wiecznie, po nas przyjdą następne ekipy rządzące. Potrzebne jest skumulowanie wiedzy, ciągłość tych polityk po to, by każdy kolejny rząd nie wynajdował koła od nowa i by nie było takiego koncertu życzeń, jaki tu dzisiaj słyszeliśmy: a może zróbmy to, a może zróbmy tamto, a może zróbmy coś innego. Potrzebne są badania, potrzebna jest polityka oparta na wiedzy. To nie jest tak, że coś, co wprowadzili Francuzi 30 lat temu, dzisiaj zadziała w Polsce, jak mówił pan poseł z Konfederacji. Polityki się rozwijają, są różne nowe odkrycia, nowe badania na świecie. Taki ośrodek powinien również służyć temu, żeby śledzić najnowsze badania światowe. A my dzisiaj, przygotowując chociażby strategię demograficzną, korzystaliśmy, szanowni państwo, z oceny, z ewaluacji programu 500+ wykonanej - przez kogo? - przez amerykańskie instytuty.

Oczywiście, że 30 mln zł można wydać na wiele innych celów, ale trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest cel dla nas istotny, czy chcemy, by polityki demograficzne w Polsce były prowadzone w spójny sposób, konsekwentnie, długofalowo, a nie chaotycznie, nie od kadencji do kadencji. Dzisiaj potrzeba nam konsekwencji, bo tylko wtedy te polityki będą skuteczne. Każdy demograf powie, że w momencie.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela wnioskodawców pana posła Bartłomieja Wróblewskiego.

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę debatę. Bardzo za niego dziękuję, ale dziękuję też wszystkim innym, którzy zabraliście dzisiaj głos.

Będę omawiał po kolei, zgodnie z tym, jak były zgłaszane różne uwagi. Do niektórych spraw już nie będę wracał, jeśli były wcześniej podniesione. Dlaczego? Dlatego że podstawy aksjologiczne tego instytutu zostały stworzone przez Platformę Obywatelską i jej poprzedników politycznych. Kto stworzył polską konstytucję?

Zwrócę też uwagę na niekonsekwencje. Z jednej strony była Unia Wolności, z drugiej strony był PSL, dalej była oczywiście Lewica, ówczesny największy klub, i Unia Pracy.

Dalej. Podpisali się pod tą konstytucją, głosowali za tą konstytucją i pan prezes, przewodniczący Tusk, i np. pan marszałek Borusewicz, i Aleksander Kwaśniewski. Krótko mówiąc, ważne osoby. Ale był w Senacie i też. Wydaje mi się, że był wicemarszałkiem, że był w Senacie. No dobrze. W każdym razie byli to politycy Unii Wolności. Padł zarzut, że prezes będzie praktycznie nieodpowiedzialny. Zwracam uwagę, pani poseł, mówię do pani poseł Rosy, że taka sama konstrukcja jest w przypadku innych rzeczników. I rzecznik praw obywatelskich, i rzecznik praw dziecka, i prezes IPN-u, i szef NBP, i szef NIK-u są praktycznie nieodpowiedzialni, ale dzięki temu mają niezależność, autonomię, mogą wykonywać działania w jakimś sensie kontrolne w stosunku do pozostałej władzy publicznej. Szef NIK-u je wykonuje, rzecznik praw obywatelskich je wykonuje, rzecznik praw dziecka je wykonuje.

Rzecznik praw obywatelskich wcześniej funkcjonował, a mimo to stworzyli instytucję rzecznika praw dziecka. Później powstawały kolejne instytucje rzeczników. Innymi słowy można powiedzieć, że ta tendencja, żeby tworzyć kolejne instytucje rzeczników, nie jest tendencją nową. Ona trwa od kliku dziesięcioleci nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Trzeba powiedzieć i oddać szacunek ministrowi Ziobrze, Ministerstwu Sprawiedliwości, że to nasze ministerstwo, nasz rząd, a później cały parlament przyjęły przepisy chroniące przed przemocą domową. Krótko mówiąc, duża rzecz w tej dziedzinie została zrobiona, a nie została zrobiona wcześniej. Pani poseł Rosa mówiła: wartości, które wam odpowiadają. Komu odpowiadały te wartości? Te wartości odpowiadały dzisiejszemu centrum, dzisiejszej lewicy.

Przechodzę do uwag pani poseł Nowickiej z Lewicy. Tutaj było dużo takich uwag ad personam, a wiemy, że uwagi personalne są najsłabszymi w każdej dyskusji. Nie będę prezesem tego instytutu. Nie zamierzam rezygnować z mandatu.

Mam prośbę do pani poseł Górskiej, żeby podała mi laptopa. Ta sprawa jest bardzo ważna.

Nie, w żaden sposób instytut nie będzie dublował pracy innych instytucji naukowo-badawczych. Natomiast w zakresie obrony praw rodziny, praw rodziców, tak jak powiedziałem, będzie w jakimś stopniu uzupełniał działanie rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka. Przechodzę do pani pytania, bardzo ważnego pytania.

Pkt 6: może zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przystępujących prokuratorowi. Czy z powodu tych przepisów pani poseł albo ktokolwiek z państwa kiedykolwiek nazywał panią rzecznik Łętowską, panów rzeczników Zielińskich, pana rzecznika Zolla, pana rzecznika Bodnara prokuratorem? To jest argument demagogiczny.

Pkt 3a: może wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich na prawach przystępujących prokuratorowi. Pkt 5: może zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przystępujących prokuratorowi. Innymi słowy, te regulacje obowiązują w Polsce od kilkudziesięciu lat.

Siłą rzeczy te przepisy dotyczące instytutu rodziny i demografii w tym zakresie, w którym ma bronić praw, konstytucyjnych praw rodziny, są analogicznie ukształtowane. To jest to, co w Polsce od dawna obowiązuje. Pojawiał się wielokrotnie zarzut, rozpoczynając już od pani poseł Nowickiej, że instytut będzie komuś kreował życie. Nie będzie nikomu kreował życia, bo w ogóle to nie jest obszar jego działalności. Jest instytucją, która ma badać, która ma analizować, która ma proponować, która ma promować rodzinę, natomiast nikogo do niczego zmuszać nie będzie. Przechodzę do uwag pani poseł Żelazowskiej, do stanowiska Koalicji Polskiej. Jest prawdą, że będzie to kolejna instytucja publiczna.

Pytanie, czy ten cel, jakim jest nawet nie zmiana trendów cywilizacyjnych, bo to jest niemożliwe, ale osłabienie tych trendów, zwiększenie przyrostu naturalnego, dzietności kobiet chociaż o jedną dziesiątą, dwie dziesiąte, trzy dziesiąte.

Jest to pewien koszt, ale w stosunku do tego, jaka jest stawka, jest to koszt naprawdę niewielki.

Czy nie lepiej pomóc ministerstwu rodziny? Instytut ma powstać po to, żeby pomagać rządowi, parlamentowi w kreowaniu polityki demograficznej, ale jednocześnie nie ma być instytucją, która jest na zawołanie parlamentu czy rządu.

Nawet jeden z departamentów ma taką nazwę: współpracy z samorządami. Pani poseł Żelazowska wspomniała o wydłużeniu urlopów macierzyńskich dzięki Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Też często powtarzam, że to była dobra rzecz, którą udało się zrobić poprzednim parlamentom. Chciałbym, żeby dzisiejsza opozycja też rozumiała, że wiele rzeczy nie ma służyć PiS-owi, tylko jest po prostu dobrymi rzeczami, które robimy w Polsce, które mają trwać przez lata, przez dziesięciolecia. Sprawdziłem to w międzyczasie. W 2015 r. na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wydawaliśmy w Polsce 170 mln zł.

Mam inne pytanie: Czy stać nas na to, żebyśmy przez kolejne lata i dziesięciolecia nic nie zrobili w sprawie demografii? Nie stać nas, proszę państwa. Nie chcę czynić zarzutów poprzednim rządom, chociaż słusznie zostało powiedziane, że przecież problem demograficzny nie powstał w ostatnich latach. Czy w wystąpieniu, formułując uzasadnienie, obciążałem rządy Platformy Obywatelskiej? Czy obciążałem lewicę? Nie obciążałem, dlatego że wszyscy rozumiemy, że problem demografii to problem cywilizacyjny, który dotyka wszystkie państwa europejskie - w różnym stopniu, ale wszystkie. Krótko mówiąc, trudno się wzajemnie przerzucać winą. To nie ma żadnego sensu. Szanowny Kolego Sośnierz z Konfederacji! Przytoczę pewne doświadczenie.

Przecież to jest niezgodne z takim klasycznym wolnościowym, liberalnym założeniem. Powiedział: W zasadzie masz rację, ale biorąc pod uwagę skalę ingerencji władzy europejskiej, rządowej, samorządowej w działalność gospodarczą, taka instytucja jest potrzebna, ponieważ przeciętny przedsiębiorca nie jest w stanie sobie poradzić. Musimy mieć taką instytucję.

Bardzo dziękuję. Krótko mówiąc: moja odpowiedź jest taka jak pana prezesa Kaźmierczaka. Rozumiem ten zarzut, w jakimś sensie zawsze stawiam to samo pytanie, co pan dzisiaj, ale uważam, że sprawa jest fundamentalna dla naszej przyszłości. Zgadzam się z wieloma takimi obserwacjami historycznymi, ale uważam, że dzisiaj nie możemy zostawiać tej sprawy własnemu biegowi. Powinniśmy zrobić to, co możemy. Padły bardzo nieeleganckie słowa ze strony pani poseł z Polski 2050.

Nikogo instytut zastraszać nie będzie. Nie jest to największa potrzeba, ale jest to rzecz jedna z wielu potrzebnych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, to, że program 500+ kosztuje ponad 30 mld zł rocznie, to 30 mln zł na instytut nie jest, wydaje się, jakimś wydatkiem bardzo dużym. W Polskim Ładzie podwyższamy kwotę wolną od podatku, a więc obniżamy podatki. Duże rodziny nie będą płacić PIT. Pani poseł. Pani marszałek. Przepraszam.

Bardzo proszę, jeszcze ma pan 2 minuty. Dobrze. Większość argumentów i kwestii została już poruszona. Padł zarzut, że po 2015 r. demografia nie skoczyła do góry, ale jednak według badań GUS w 2020 r. dzietność w Polsce miała wynosić 1,28 dziecka na kobietę, natomiast dane pokazują, że jest to 1,41, czyli, krótko mówiąc, został zahamowany spadek przyrostu naturalnego w Polsce. Moim zdaniem taki powinien być właśnie cel instytutu. Prawdą jest to, co powiedział pan poseł Woźniak, że dla niektórych uczestników tej dyskusji jest to kolejna okazja do tego, żeby zaatakować rodzinę.

Nie będzie żadnego nepotyzmu. Celem instytutu jest stworzenie instytucji merytorycznej. Zarówno prezes, jak i członkowie rady, ale także pracownicy muszą się wykazać odpowiednimi kompetencjami w zakresie wiedzy o rodzinie, demografii, w zakresie prawa, żeby mogli znaleźć zatrudnienie w instytucie.

Mogę powiedzieć, że projekt jest gotowy. Mam nadzieję, że wkrótce będzie decyzja polityczna i ten projekt trafi do Sejmu. Uważam, że sprawa jest ważna, też mi na tym zależy, i myślę, że większości Wysokiej Izby na tym zależy. Pani poseł Skowrońska, bardzo proszę o spokój. Panie pośle, bardzo proszę zbliżać się do końca.

Jeszcze raz: po pierwsze, rzetelna praca analityczna, rzetelna praca naukowa związana ze sprawami rodziny, z polityką demograficzną, po drugie, tworzenie propozycji polityk w zakresie rodziny, w zakresie demografii, po trzecie, promocja rodziny, prowadzenie programów społecznych, które zachęcą Polaków do posiadania dzieci, tworzenia rodzin, które będą tworzyły przyjazny klimat rodziny, i po czwarte, obrona konstytucyjnych wolności i praw, które zostały zapisane w konstytucji, w taki sposób, jaki został zapisany w konstytucji.

Dziękuję, panie pośle. Zgadzam się, że konstytucja jest bardzo ważna i należy jej przestrzegać we wszystkich punktach. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań.

Jeżeli nie, to zamykam listę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Wojenną, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Podpisano naczelnik państwa Józef Piłsudski. Ów dekret, tworząc formalnie marynarkę wojenną, miał doniosłe konsekwencje, wydany w warunkach, kiedy tylko niewielka część ziem polskich była w naszych rękach i płonęły właściwie wszystkie granice. Pomorze pozostawało w niemieckich rękach, a jego odzyskanie wydawało się jeszcze wtedy mało prawdopodobne. Akt wyraźnie artykułował polskie prawa dostępu do morza, podkreślał także polskie roszczenia wobec Gdańska. Jej zręby, co oczywiste, tworzyli oficerowie i marynarze służący kiedyś we flotach państw zaborczych. Pierwszą bazą był port rzeczny w Modlinie, a zanim polscy marynarze wpłynęli na ołowiane fale Bałtyku, zdali bojowy egzamin, walcząc na rzekach i jeziorach w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Pierwszym bojem polskiej floty była stoczona w kwietniu 1920 r. bitwa pod Czarnobylem, kiedy to polskie okręty zniszczyły kilka sowieckich jednostek. Wisły przed oskrzydlającymi wojskami sowieckimi. Wielu z nich zostało odznaczonych Orderem Virtuti Militari. Kiedy w końcu uzyskano dostęp do morza, na tym naszym skrawku Wybrzeża zaczęto się bardzo pracowicie krzątać i przygotowywać flotę. Przyznanych nam przez sojusznicze rady ambasadorów kilka niewielkich okrętów nie zaspokoiło polskiego apetytu. Niestety możliwości finansowe zniszczonego przez wojnę, tworzonego na nowo państwa sprowadzały na ziemię tych, którzy widzieli Polskę jako potęgę na morzu.

Znalazły się w niej zarówno nowoczesne, jeśli nie najnowocześniejsze, kontrtorpedowce na Bałtyku typu „Grom”, dwa typu „Wicher”, pięć okrętów podwodnych, w tym dwa oceaniczne „Sęp” i słynny „Orzeł”, kilka trałowców i stawiaczy min. W kampanii wrześniowej młoda flota zdała egzamin, mimo że część okrętów ewakuowano do Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy wydzierżawili PWM kilkanaście jednostek, na których polscy marynarze dokonywali cudów waleczności.

Po roku 1945 warunki zmieniły się całkowicie. Polska otrzymała ogromny obszar wybrzeża Bałtyku, który wymagał ochrony.

Ochrona naszego Wybrzeża jest kluczowa dla niepodległości Polski. Rozbudowa Marynarki Wojennej jest elementarna dla bezpieczeństwa naszego państwa. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, ale w szczególności pracowników socjalnych. Czym się zajmują pracownicy socjalni? Pomagają osobom i ich rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Wspierają beneficjentów pomocy społecznej w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Dużo czasu i uwagi poświęcają pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Współuczestniczą w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Aby pracownik socjalny mógł sprawnie wykonywać swoje zadania, musi spełniać wiele wymogów, które formułuje ustawa o pomocy społecznej. Chodzi tu z jednej strony o odpowiednie specjalistyczne wykształcenie zdobyte w kolegium dla pracowników służby społecznych, na studiach na kierunku praca socjalna lub na innym kierunku w tym zakresie, a z drugiej - o dwustopniową specjalizację zawodową. Obecnie w ośrodkach społecznych i w powiatowych centrach pomocy rodzinie pracuje ponad 20 tys. pracowników socjalnych. Dzięki działaniom pracowników socjalnych wiele osób staje na nogi i zmienia swoje życie. Pracownicy socjalni to bohaterowie, którzy nie noszą peleryn. Wykonywanie ich zawodu nierzadko wiąże się z narażeniem zdrowia lub życia. Wszystkim pracownikom socjalnym z okazji ich święta składam serdeczne życzenia zdrowia, dużo sił na każdy dzień, wyrozumiałości dla innych, satysfakcji z wykonywanej pracy. Pan poseł Bartłomiej Dorywalski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Pacyfikacja Kurzelowa.

W tym dniu niemiecka żandarmeria z Włoszczowy i Kluczewska otoczyła Kurzelów i rozpoczęła się jego pacyfikacja. Ok. 60 mężczyzn zostało wprowadzonych ze swoich domów i zebranych przed budynkiem nadleśnictwa. Mężczyźni, którzy stawiali opór, byli eliminowani w miejscu zatrzymania. Już w tym czasie podczas zatrzymania zastrzelono dwie osoby, które próbowały uciec - Tadeusza Szczuckiego i Franciszka Czaińskiego, który zginął wyprowadzany ze swojego sklepu. Ci, którzy zostali doprowadzeni na przesłuchanie, pojedynczo wchodzili do budynku nadleśnictwa. Podczas przesłuchań dochodziło do aktów przemocy.

Po zakończeniu przesłuchań 18 mężczyzn przeprowadzono do piaskowni koło cmentarza, to tam zostali zamordowani. Odjeżdżając, Niemcy zabrali ze sobą czterech aresztowanych: Feliksa Gradońskiego ps. Spokojny, Stanisława Gieronia, Adama Stępniewicza i Antoniego Celebańskiego. Spośród 20 zamordowanych tego dnia 19 osób zostało pochowanych w dwóch mogiłach obok siebie w miejscu egzekucji na tzw. małym cmentarzu. Wiedza na temat ofiar jest bardzo uboga. Księgi parafialne, które zawierają wpisy o tragicznej śmierci, zostały sporządzone dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Panuje przekonanie, że zbrodnia ta nie doczekała się opracowania ze względu na nazwisko osoby, która sporządziła listę dla niemieckiego okupanta. Był to niemiecki agent pracujący w urzędzie gminy Kurzelów. Tym czynem wydał on na siebie wyrok śmierci i został zlikwidowany w nocy z 18 na 19 marca w momencie opanowania Włoszczowy przez oddziały Armii Krajowej. Ofiary pacyfikacji Kurzelowa w obliczu wojny i stałego zagrożenia stały murem za ruchem oporu i obrońcami ojczyzny. W chwili obecnej to my jesteśmy zobowiązani stać murem za polskim mundurem, obrońcami naszych granic. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Dariusz Bąk, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. Pan poseł Władysław Kurowski, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Dziś, dbając o pamięć historyczną, chciałbym przedstawić ważne, choć tragiczne wydarzenie z powiatu myślenickiego, z gminy Tokarnia z 29 listopada 1944 r. i 4 grudnia tegoż samego roku. Wzmożone działania zbrojne wymierzone przeciwko oddziałom partyzanckim na terenie powiatu myślenickiego realizowane były przez okupanta niemieckiego od lata 1944 r. Było to spowodowane przede wszystkim działaniami operacyjnymi oddziałów partyzanckich. W odpowiedzi na te działania oraz w trosce o zabezpieczenie własnego zaplecza przed zbliżającym się frontem Niemcy podjęli radykalne i krwawe działania polegające na likwidacji zgrupowań partyzanckich.

Oddziały hitlerowskie liczyły ponad 3 tys. doskonale uzbrojonych ludzi: broń maszynowa, granatniki, moździerze, zwiad lotniczy. Przeciwko nim do walki stanęło niespełna 300 partyzantów słabo uzbrojonych. Pomimo przewagi liczebnej, ogniowej oraz zaskoczenia nie udało się Niemcom osiągnąć zakładanych rezultatów, bowiem bohaterska postawa oddziału Bicza Żelbet II zaalarmowała i dała czas na przygotowanie obrony pozostałym oddziałom partyzanckim. W pewnym momencie rozpoczęli nawet w gęstej mgle zaciętą walkę między sobą, co zwiększyło ich straty. Według strony niemieckiej poległo dziewięciu policjantów, w tym dwóch podoficerów, i siedmiu odniosło rany. Natomiast Polacy na podstawie informacji wywiadu oraz sprawozdań oddziałów terenowych Armii Krajowej ocenili straty na kilkakrotnie większe - kilkudziesięciu zabitych i rannych. Niestety na roli Tajsowej przed południem 29 listopada 1944 r. ginęli również cywilni mieszkańcy Zawadki. Zginęło trzech mężczyzn bezpośrednio od strzału w tył głowy. Natomiast Aniela Mizera i Andrzej Tajs zginęli od zabłąkanych kul i następnie spalili się w ich płonących domostwach. Andrzej Kowalik z roli Jaworzyny został ciężko pobity i w efekcie poniesionych obrażeń zmarł. W tym miejscu należy również wspomnieć anonimowego mieszkańca Krzczonowa, który został skatowany do nieprzytomności za to, że prowadził Niemca w stronę Zawadki zbyt opieszale i nie najkrótszą drogą. Jan Rapacz zabrany w dniu 4 grudnia przez Niemców z Zawadki zaginął bez wieści, prawdopodobnie został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Żołnierze Żelbetu polegli w walce oraz Andrzej Kowalik z Jaworzyny zostali następnego dnia przetransportowani na cmentarz parafialny w Trzebuni i tam pochowani. Ciała żołnierzy po wojnie zostały ekshumowane i przewiezione na cmentarz Rakowicki w Krakowie. Pozostałe ofiary pacyfikacji Zawadki w nocy 29 listopada zostały pochowane we wspólnej mogile na cmentarzu w Krzczonowie z inicjatywy dowódcy partyzanckiego oddziału dywersyjnego Franciszka Pytlika, który przygotował transport ciał pomordowanych i trumny do pochówku. Niestety już po kilku dniach, bo już 4 grudnia 1944 r., na kilka godzin przed świtem z Myślenic i Krakowa wyruszyła karna ekspedycja udająca się w rejon masywu Kotonia z zamiarem ukarania mieszkańców, którzy pomagali partyzantom, oraz zlikwidowania potencjalnej bazy partyzanckiej. Penetrowano również teren w poszukiwaniu zaginionych Niemców. Okupant hitlerowski, stosując bezwzględną zasadę zbiorowej odpowiedzialności, mścił się na bezbronnej ludności cywilnej, która zapłaciła ogromną cenę za to, że Zawadka stała się bazą partyzancką. Spalone zostały wszystkie zabudowania. Niemcy swoich barbarzyńskich działań nie ograniczali tylko do Zawadki, spalili również domy w sąsiednich wsiach. W Zawadce zostały tylko przydrożne kamienne kapliczki i krzyże oraz drewniana kuźnia. W Pcimiu okupant spalił kilkanaście gospodarstw na różnych rolach. Wszyscy mieszkańcy ocaleni z pożogi, bez jakichkolwiek środków do życia, na czas mroźnej i śnieżnej zimy schronili się u swoich krewnych i znajomych w okolicznych wsiach. Po wojnie w 1964 r. z inicjatywy żołnierzy Armii Krajowej i przy współpracy władzy gminnej na roli Tajsowej w Zawadce wybudowano kamienny obelisk, a na nim wmurowano dwie tablice upamiętniające zbrojny czyn polskiego podziemia oraz tragiczną śmierć mieszkańców. Co roku we wrześniu w tym miejscu sprawowana jest msza święta i odbywają się uroczystości upamiętniające walki w masywie górskim Kotonia i tragiczną pacyfikację Zawadki. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Pieczęć Zasług Obywatelskich przyznawana jest od 2016 r. To honorowe odznaczenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, które otrzymują mielczanie wybitnie zasłużeni dla ziemi mieleckiej oraz dla ojczyzny. W przeszłości byli to m.in. odznaczeni pośmiertnie bł. ks. Roman Sitko, prof. Władysław Szafer - urodzony na ziemi mieleckiej, gen. broni Władysław Sikorski, bracia Działowscy - Stanisław i Mieczysław, prekursorzy mieleckiego i polskiego lotnictwa, oraz żyjący współcześnie m.in. były prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski, konstruktor lotniczy Józef Oleksiak czy ks. prałat Kazimierz Czesak.

Andrzej Kędzior, o którym krótko można powiedzieć, że ratował przed głodem i powodziami, urodził się 7 listopada 1851 r. w Toporowie pod Mielcem. Rodziców nie było stać na finansowanie synowi nauki w gimnazjum, dlatego syn, wybitnie uzdolniony, zarabiał jako korepetytor zamożnych kolegów, których rodzice pomogli mu studiować w Wiedniu - najpierw na politechnice, potem meliorację na akademii rolniczej, a następnie także prawo na uniwersytecie. Po ukończeniu nauki w 1879 r. otrzymał posadę inżyniera w utworzonym właśnie Krajowym Biurze Melioracyjnym we Lwowie. Andrzej Kędzior osobiście napisał austriacką ustawę wodną, przyjętą w 1884 r. Za sprawą jego i jego współpracowników obwałowano rzeki i odwodniono rolnicze użytki niziny krakowsko-sandomierskiej i Doliny Nadwiślańskiej powyżej Krakowa, a także obszary w dorzeczu Dniestru, górnego Bugu, Styru. Wały zabezpieczające po dziś dzień przed wylewem Wisły, Rudawy, Raby, Dunajca, Brnia, Trzęsówki, Sanu oraz niezliczonych odcinków innych cieków wodnych są jeśli nie bezpośrednim dziełem koncepcyjnym inżyniera spod Mielca, to powstały według nakreślonych przez niego planów bądź projektów.

Był również inicjatorem budowy kanału Wisła-Odra-Dniestr, a także sprawował m.in. funkcję ministra robót publicznych w polskim rządzie Jędrzeja Moraczewskiego i Leopolda Skulskiego.

Został odznaczony również Orderem Polonia Restituta z gwiazdą. Spoczął na cmentarzu w Mielcu. Kolejnym tegorocznym laureatem odznaczonym Pieczęcią Zasług Obywatelskich jest pan Józef Witek - wybitny znawca regionu, kronikarz, animator kultury, społecznik, autor książek dotyczących historii Mielca i ziemi mieleckiej, w tym m.in. 4-tomowej Encyklopedii Miasta Mielca. Józef Witek jest rodowitym mielczaninem. Przez wiele lat był choreografem i instruktorem zespołów tanecznych i muzycznych. To już kilkanaście różnych pozycji, m.in. o ulicach i ich patronach, jak również publikacje poświęcone (Dzwonek) m.in. szkole muzycznej czy Stali Mielec. Ale najwięcej pracy kosztowało go stworzenie Encyklopedii Miasta Mielca. W swojej książce regionalista umieścił wiele tysięcy haseł. Oprócz biogramów ludzi są informacje o ulicach i placach, hasła geograficzne, przyrodnicze, przemysłowe, handlowe, komunalne czy urzędnicze, a więc wszystko, co składa się na życie miasta. Podczas uroczystości wręczenia Pieczęci Zasług Obywatelskich wręczono również odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane panu Piotrowi Pszenicznemu - wyróżniającemu się artyście malarzowi i rzeźbiarzowi, członkowi Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej z okazji 40-lecia klubu. Wszystkim odznaczonym składam serdeczne gratulacje, a Towarzystwu Miłośników Ziemi Mieleckiej dziękuję za piękną inicjatywę zatrzymywania mijającego czasu. Chcę jeszcze również poinformować szanownych państwa o jubileuszu 75-lecia Teatru Rozmaitości im. Stefana Ostrowskiego w Mielcu, jedynego w swoim rodzaju teatru amatorskiego wystawiającego różnego rodzaju spektakle.

Gratuluję artystom i życzę dalszych sukcesów. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie!

Do sprzysiężenia przystąpiło ok. 200 członków. Przez kilkanaście miesięcy przygotowywano się do wystąpienia zbrojnego. Rok 1830 przyniósł w Królestwie Polskim radykalizację nastrojów wynikającą z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej będącej wynikiem wzrostu cen żywności i pojawiającego się bezrobocia. W Warszawie dochodziło do spontanicznych strajków, a nawet drobnych rozruchów. W lipcu 1830 r. wybuchła rewolucja we Francji, w wyniku której obalono Burbonów, a w sierpniu Belgowie rozpoczęli walkę o niepodległość, której celem było oderwanie się od Holandii. Ogłoszony 19 i 20 listopada 1830 r. rozkaz stawiający w stan pogotowia armię rosyjską i Wojsko Polskie wierne carowi jako królowi polskiemu zmusiło Piotra Wysockiego i pozostałych spiskowców do podjęcia natychmiastowych działań. Termin wybuchu powstania zbrojnego wyznaczono na dzień 29 listopada 1830 r. na godz. 18. W tym czasie w Warszawie stacjonowało ok. 6,5 tys. żołnierzy rosyjskich i ok. 10 tys. żołnierzy polskich. O godz. 18. podpalono browar na Solcu, co miało być sygnałem do jednoczesnego rozpoczęcia wszystkich działań zbrojnych. Piotr Wysocki poderwał do broni ponad 160 podchorążych. Liczono na pozyskanie mieszkańców Starego Miasta i większości oddziałów Wojska Polskiego pozostających dotychczas pod komendą wielkiego księcia Konstantego. Niechęć do przyłączenia się do insurekcji kolejnych generałów cieszących się uznaniem powstańców skutkowała tym, że kilku z nich zabito. Obawy znacznej części mieszkańców stolicy, którzy po prostu bali się wojny i ewentualnych represji, też nie rokowały dobrze w pierwszych godzinach zrywu. Mimo to w ciągu nocy powstańcy opanowali całą Warszawę. Wielki książę Konstanty nie zdecydował się na szturmowanie stolicy, a wierne sobie oddziały wycofał do Wierzbna. W gronie powstańców podobnie jak wśród ludu w stolicy zaczęły ścierać się frakcje zwolenników otwartej walki z Rosją z konserwatystami, czyli zwolennikami negocjacji i porozumień z carem jako królem. Przeciwstawił się tym porozumieniom m.in. Joachim Lelewel, który stworzył porozumienie, stworzył Klub Patriotyczny. Jednym z najaktywniejszych członków Klubu Patriotycznego był Maurycy Mochnacki, który 1 grudnia stanął na czele Towarzystwa Patriotycznego. 3 grudnia 1830 r. w wyniku nacisków Klubu Patriotycznego utworzono Rząd Tymczasowy z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim na czele. W skład rządu wszedł m.in. Joachim Lelewel. W wyniku rokowań z księciem Konstantym jednostki polskie miały wrócić do Warszawy, zaś wojska rosyjskie na czele z samym księciem miały odejść w stronę granicy. Car nie godził się jednak na żadne ustępstwa. Powstanie przerodziło się w wojnę polsko-rosyjską. Sejm zatrzymał władzę zwierzchnią w państwie i powołał Rząd Narodowy z Adamem Jerzym Czartoryskim na czele. Rozpoczęła się wojna Polaków z przeważającymi siłami wroga. Formalnego aktu kapitulacji nigdy nie podpisano. Powstanie listopadowe jest żywe w pamięci Polaków do dnia dzisiejszego. Należy oddać hołd wszystkim powstańcom narodowym, w tym szczególnie w kolejną rocznicę wybuchu powstania listopadowego, i tym, którzy walczyli z przeważającymi siłami wroga w wojnie z Rosją w roku 1831. W roku, w którym Polska przez wiele miesięcy była de facto państwem niepodległym. Potem przyszedł czas na niemiłosierne represje wobec Polski i Polaków, ale to już temat na inne wystąpienie. Na zakończenie mojego oświadczenia pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powrotu do Polski doczesnych szczątków Maurycego Mochnackiego, bohatera tamtych czasów, który wreszcie spoczął w polskiej ziemi, w ziemi Polski niepodległej, a więc takiej, o jakiej marzył i o jaką walczył. Cześć pamięci wszystkich, którzy chwycili za broń i którzy prowadzili różnorakie działania na rzecz niepodległości Polski.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie pragnę serdecznie podziękować za dbanie o polskie dzieła sztuki, za odkupowanie cennych dla naszego narodu kolekcji i dzieł. Stają się one naszą nie tylko duchową, ale też i rzeczywistą własnością. Przyjmowanie dóbr artystycznych w ten sposób świadczy o głębokim zainteresowaniu budowaniem trwałej tożsamości narodowej. Najbardziej spektakularnym przykładem dbałości o polskie kolekcje jest odkupienie od Fundacji Książąt Czartoryskich dzieł sztuki, wśród których znajdują się m.in. obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta czy Renoira. Jak wiemy, zostały one przekazane do Muzeum Narodowego w Krakowie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera także zakupy dzieł sztuki zrabowanych w czasie zawieruchy wojennej czy zaginionych w rozmaitych okolicznościach, a także obrazów dla placówek muzealnych mieszczących się nie tylko w metropoliach, ale i w mniejszych ośrodkach.

Jako reprezentantka miasta określanego polską perłą renesansu chcę za to bardzo podziękować. Tematem „Panoramy Siedmiogrodzkiej” jest zwycięska bitwa o stolicę Siedmiogrodu rozegrana 11 marca 1849 r. pod dowództwem bohatera dwóch narodów, wywodzącego się właśnie z Tarnowa generała Józefa Bema. Muzeum Okręgowe w Tarnowie jest już właścicielem 24 spośród 60 fragmentów „Panoramy Siedmiogrodzkiej” Są one eksponowane w niezwykle ciekawym i historycznym miejscu, w Galerii „Panorama” mieszczącej się w budynku dworca kolejowego w Tarnowie. Pozyskany ostatnio fragment w pierwszych dniach grudnia także będzie można podziwiać w tym miejscu. Cieszy to tym bardziej, że Tarnów jest bodaj najbardziej węgierskim ze wszystkich polskich miast. Związki polsko-węgierskie w Tarnowie mają wielowiekową tradycję.

Chlubnie zapisało się tu przede wszystkim nazwisko gen. Józefa Bema urodzonego, jak już wspomniałam, właśnie w Tarnowie i w tym mieście pochowanego. Nie wszyscy wiedzą, że w Tarnowie w 1948 r. miały miejsce ogólnopolskie obchody 100. rocznicy Wiosny Ludów. Także tutaj przed kilkoma laty zorganizowano międzynarodowe dni przyjaźni polsko-węgierskiej. Miasto Tarnów oraz większość gmin w regionie tarnowskim posiada miasta partnerskie na Węgrzech. W centrum Tarnowa i obok podtarnowskich Koszyc Wielkich znajdują się oryginalne bramy seklerskie wykonane przez cieśli z Siedmiogrodu. Jest ich w Polsce trzy - prócz Tarnowa także w Starym Sączu. Kończąc zaproszeniem do pięknego Tarnowa, raz jeszcze dziękuję za finansowe wsparcie zakupu kolejnego fragmentu dzieła Jana Styki pod nazwą „Panorama Siedmiogrodzka” Jest ono, podobnie jak cała kolekcja, niejako wspomnianą na wstępie własnością całego naszego narodu. Muzeum okręgowe w Tarnowie nie ustaje w poszukiwaniach kolejnych fragmentów, a w planach jest także stworzenie całej ekspozycji, która byłaby jedyną taką w skali kraju i pełniłaby rolę unikatu, jakim jest np. muzeum Panorama Racławicka we Wrocławiu. Bardzo proszę, pan poseł Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pierwszy etap remontu zabytkowego mostu w Tczewie został zrealizowany za rządów PO-PSL. Od lipca 2015 r. trwa remont tego mostu, a ostatni etap prac IIA rozpoczął się w 2019 r. i cisza. Wtedy nawet prezydent Duda w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że wesprze remont tego mostu.

Niestety 30 września 2019 r. wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał prace, a środki, które starostwo zarezerwowało na dokończenie etapu IIA, musiały trafić na zabezpieczenie placu budowy przed zimą. To ok. 10 mln zł. To jest kwota nie do udźwignięcia przez powiat tczewski. Niestety posłowie PiS, nawet ci z Pomorza, z tego regionu, nie poparli przyznania pieniędzy dla starostwa tczewskiego. A tyle pięknych słów padało, że będą pracować dla dobra mieszkańców. Powiatu nie stać nawet na wkład własny, który jest niezbędny przy dofinansowaniu ze środków rządowych. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana właściciela mostu, dlatego starostwo powiatowe w Tczewie od lat apeluje o przejęcie mostu przez Skarb Państwa - bezskutecznie. W tym celu napisałam nawet projekt ustawy przejęcia tego mostu przez Skarb Państwa jako oddziału Muzeum II Wojny Światowej. Przecież na tym moście rozpoczęła się II wojna światowa. Ostatnio dodatkowo starostwo powiatowe w Tczewie złożyło wniosek do rządowego programu inwestycji lokalnych w ramach Polskiego Ładu o sfinansowanie aktualizacji projektu budowlanego remontu mostu. Rząd przyznał 684 tys.

Zwracam uwagę, przypominam, że wojewódzki konserwator zabytków został powołany przez PiS. Apeluję więc po raz kolejny z tej mównicy do rządu o jak najszybsze przejęcie mostu tczewskiego przez Skarb Państwa i jego szybką odbudowę. Most ten to nie tylko wspaniały zabytek architektury inżynieryjnej XIX w., ale też ważna trasa komunikacyjna dla mieszkańców między Tczewem a Lisewem Malborskim. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Maria Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. Pan poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Adam Chmielowski to polski zakonnik franciszkański, założyciel zgromadzeń albertynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty Kościoła katolickiego. Znany z pełnej poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych. To postać znana oczywiście w całej Polsce, ale też szczególna dla mojego miasta, dla Puław.

Misją towarzystwa jest skupianie ludzi dobrej woli, pragnących działać dla dobra drugiego człowieka w duchu swojego patrona poprzez tworzenie schronisk, noclegowni, łaźni, kuchni, z których korzystają ludzie potrzebujący pomocy. Od początku istnienia schroniska w Puławach udzielono schronienia tysiącom osób, a wielu innym pomocy doraźnej w formie posiłku, odzieży lub pojedynczego noclegu. Koło towarzystwa prowadzi też działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans i w zakresie ochrony zdrowia, poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Schronisko przeznaczone dla mężczyzn posiada ok. 40 miejsc stacjonarnych, w okresie zimy w razie potrzeby ta liczba jest zwiększana. Zapewnia schronienie, całodzienne wyżywienie, kąpiel, wymianę odzieży, systematyczną opiekę duszpasterską, kontakty z poradnią odwykową oraz pomoc socjalną.

W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości, wyrażających w swoich wystąpieniach szacunek i uznanie dla dokonań towarzystwa i dziękujących kierownictwu oraz wszystkim członkom zaangażowanym w działalność. Duża grupa pracowników koła została wyróżniona stosownymi odznakami lub dyplomami. Pracownicy ci to jedna wielka rodzina osób poświęcających się pomocy potrzebującym bliźnim, ludziom ubogim, nieradzącym sobie z trudnościami codziennego życia, bezdomnym żyjącym w oderwaniu od rodzin. Kierownictwu i członkom Puławskiego Koła Towarzystwa z okazji jubileuszu 30-lecia składam serdeczne gratulacje i podziękowania. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W kończącym się miesiącu listopadzie br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy obchodziła 10. rocznicę nadania imienia Mariana Rejewskiego. Ten znakomity bydgoszczanin, wybitny matematyk, genialny kryptolog złamał niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Dokonanie tego miało ogromny wpływ na losy II wojny światowej. Bardziej przyczynił się do zwycięstwa aliantów nad Hitlerem niż wszystkie armie, napisał o nim Jan Nowak-Jeziorański.

Polacy przekazali aliantom i podzielili się informacjami, jak łamać szyfr Enigmy. Dlatego warto przedstawić tę wyjątkową placówkę, która swoimi dokonaniami angażuje się w promowanie edukacji historycznej, obywatelskiej i regionalnej. Początki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i jej zbiorów sięgają roku 1921, kiedy to powstała Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. Kolejne losy sprawiały, że biblioteka zmieniała swoje siedziby i lokalizację, by ostatecznie od roku 1968 wrosnąć w edukacyjną przestrzeń Bydgoszczy. Od ponad 50 lat biblioteka stanowi jedną z najbardziej aktywnych i znaczących instytucji w regionie, ze zbiorami na poziomie 173 tys. jednostek inwentarzowych. Systematycznie rozbudowuje księgozbiór wydawnictw pedagogicznych i psychologicznych oraz socjologicznych. Jej bogate zbiory, w tym archiwalia i muzealia gromadzone w Muzeum Oświaty, które wchodzi w strukturę tej placówki, jak i wszelkie usługi dostępne są dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu. Biblioteka systematycznie modyfikuje i podnosi atrakcyjność oferty edukacyjno-kulturalnej. Kontynuuje i rozwija kilka projektów oświatowych oraz proponuje bogaty zestaw zajęć edukacyjnych. Z urozmaiconej oferty biblioteki mogą korzystać wszystkie grupy odbiorców, poczynając od najmłodszych poprzez uczniów, studentów, nauczycieli po seniorów. Jednak najważniejszy jest fakt, że swoje działania wychowawcze biblioteka oparła na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Mariana Rejewskiego, dla którego najważniejsze było dobro ojczyzny. Dlatego od 10 lat Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy popularyzuje zasługi swego patrona w regionie i w Polsce, przywracając Marianowi Rejewskiemu i polskim kryptologom właściwe miejsce w historii Polski i świata. Od czasu przyjęcia imienia biblioteka realizuje projekt edukacyjny pod nazwą: Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog. W lekcjach o Marianie Rejewskim wzięło udział ponad 7 tys. uczniów. Wystawę pod tym samym tytułem w większych i mniejszych miastach województwa kujawsko-pomorskiego odwiedziło ok. 15 tys. uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców. Biblioteka aktywnie angażuje się w upowszechnianie pamięci historycznej i budowanie własnej tożsamości młodego pokolenia. Różnorodne i innowacyjne formy edukacyjne rozwijają kompetencje i zainteresowania matematyczne, umiejętności intelektualne i społeczne, wspierają także działania dydaktyczne szkół i nauczycieli.

Organizuje wystawy, konferencje, seminaria, warsztaty i konkursy. Od wielu lat mam zaszczyt obserwować dokonania i rozwój tej instytucji. Biblioteka ta jest placówką dbającą o wysoką jakość świadczonych usług, promującą wartość uczenia i doskonalenia przez całe życie. Służy kształcącym i doskonalącym się nauczycielom oraz studentom przygotowującym się do wykonywania zawodu. Z okazji jubileuszu nadania imienia życzę pedagogicznej bibliotece w Bydgoszczy stałego rozwoju pod względem zasobów bibliotecznych, infrastruktury, a kadrze nauczycielskiej życzę, by właściwie wypełniała swoją misję cenionego ośrodka informacji oświatowej, regionalnej i kulturalnej. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Samorządowcy z Ziemi Lubuskiej! Zechciejcie nakłonić ucha, bo chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, co było moim udziałem w ostatnim tygodniu. Tak się składa, że poselska mitręga ma swoje odzwierciedlenie nie tylko tutaj, na sali parlamentarnej Wysokiej Izby, ale również w okręgu, gdzie realizujemy pracę organiczną na rzecz naszych regionów, w moim przypadku ziemi lubuskiej. Zatem ostatni tydzień to był cykl spotkań z samorządowcami z jednostek samorządu terytorialnego, do których pojechałem, by ponownie podyskutować o kolejnym etapie przygotowywania projektów w ramach programu Polski Ład.